Wznawiam obrady. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 2. porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Przypominam, że postawienie pytania nie może trwać dłużej niż 2 minuty, zaś udzielenie odpowiedzi nie może trwać dłużej niż 5 minut. Prawo do postawienia pytania dodatkowego przysługuje wyłącznie posłowi zadającemu pytanie. Dodatkowe pytanie nie może trwać dłużej niż 1 minutę, a uzupełniająca odpowiedź nie może trwać dłużej niż 3 minuty. Marszałek Sejmu może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu odpowiedzi na pytanie dodatkowe.

Pytanie jest w sprawie rozwoju jednostek ochotniczych straży pożarnych i rządowego wsparcia dla jednostek OSP na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Pytanie jest skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji. Bardzo proszę, pani poseł Joanna Borowiak.

Bardzo proszę. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Ochotnicza straż pożarna to bardzo ważne skrzydło ochrony przeciwpożarowej w Polsce, a lokalne jednostki OSP są swoistym buforem bezpieczeństwa dla mieszkańców społeczności, w których funkcjonują. Strażacy ochotnicy są zawsze we właściwym miejscu i właściwym czasie, gotowi nieść pomoc przy gaszeniu pożarów, ratować ludzkie życie i mienie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w zakresie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, doposażenia jednostek, przekazywania środków finansowych na potrzebny sprzęt i remonty remiz. Opozycja już kilka razy wieszczyła koniec ochotniczej straży pożarnej za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Panie Ministrze! Jak to wygląda z dzisiejszej perspektywy? Jakie środki finansowe zostały przeznaczone na wsparcie funkcjonujących jednostek? Jakie działania zostały podjęte przez rząd, aby strażacy ochotnicy mogli nieść pomoc Bogu na chwałę, ludziom na pożytek? I jeszcze jedno: Jak strażacy, druhowie ochotnicy oceniają rządowe wsparcie? Dziękuję bardzo, pani poseł. O udzielenie odpowiedzi na pytanie bardzo proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji ministra Macieja Wąsika. Bardzo proszę, panie ministrze. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Rząd Prawa i Sprawiedliwości docenia ogromną rolę, jaką ochotnicze straże pożarne odgrywają w realizacji zadań w obszarze ochrony przeciwpożarowej. Rząd podejmuje liczne działania na rzecz podnoszenia poziomu wyposażenia i wyszkolenia tych jednostek oraz zapewnienia dofinansowania ich działalności ze środków budżetu państwa.

Wysokość środków finansowych, które trafiały do jednostek OSP, pozwalała na zauważalne podnoszenie ich standardów i wyposażenia. Podkreślenia wymaga, że pomimo iż kwoty przeznaczone dla OSP w ostatnich latach są naprawdę wysokie, nie są w stanie pokryć wszystkich niezbędnych potrzeb tych jednostek. W 2020 r., dzięki wspólnym staraniom i bardzo dobrej współpracy właściwych ministrów: do spraw klimatu i środowiska oraz spraw wewnętrznych i administracji, na podstawie porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska jednostki OSP otrzymały ogromne wsparcie finansowe ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, chodzi o kwotę 143 660 tys. zł. Na podkreślenie zasługuje fakt, że zakupy samochodów pożarniczych dla jednostek OSP w całym kraju realizowane były przez komendanta głównego PSP w ramach montażu finansowego ze środków pochodzących z różnych źródeł: z budżetu państwa, z budżetów jednostek samorządowych utrzymujących OSP, z funduszów ochrony środowiska, jak również ze źródeł pozabudżetowych, które to środki komendant główny PSP otrzymał od zakładów ubezpieczeń, a uzyskane zostały z tytułu obowiązującego ubezpieczenia od ognia.

Warto podkreślić, że kwoty te umożliwiły zakupienie dla ochotniczej straży pożarnej największej od wielu lat liczby specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Tak że można powiedzieć, że w ostatnich latach potroiła się pomoc państwa dla ochotniczych straży pożarnych.

Chciałbym jeszcze podkreślić, że z zasobów Państwowej Straży Pożarnej do jednostek OSP trafiają samochody używane, które są wycofywane, zgodnie ze standardami, które określa komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.

Oprócz tego trafia oczywiście różnego typu sprzęt.

W ten sposób wyremontowano czy zmodernizowano prawie 2700 strażnic OSP.

Mamy w tej chwili - jak ocenia komendant główny Państwowej Straży Pożarnej - ponad 200 tys. strażaków ratowników, którzy posiadają uprawnienia do udziału w działaniach ratowniczych. Bardzo dziękuję. Dziękuję, panie ministrze. Z pytaniem dodatkowym pan poseł Waldemar Andzel. Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Chciałem jeszcze dopytać, jak to będzie wyglądało w kolejnych latach. Czy nadal będzie takie wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych? Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Pan minister Maciej Wąsik. Pani Marszałek! Panie Pośle! W tym roku, pomimo ciężkiej sytuacji COVID-owej, udało się stworzyć pewną inżynierię finansową w oparciu o środki ministerstwa, w oparciu o środki narodowego funduszu i środki samorządów, z których zakupiono ponad 300 samochodów dla ochotniczych straży pożarnych. Państwowa Straż Pożarna dokonuje zakupu nowej floty, wprowadza nowe samochody do użycia. Te dotychczasowe, całkiem sprawne, to są samochody - powiedzmy - 10-, 12-, 15-letnie, dobrze utrzymane, są one przekazywane do ochotniczych straży pożarnych, w szczególności do tych, gdzie samorządy nie są w stanie wyasygnować środków na wkład własny na zakup nowych aut ratowniczo-gaśniczych. Chciałem także podkreślić, że ciągle pamiętamy, próbujemy zaplanować budżet na przyszły rok. Jestem przekonany, że rząd doceni OSP i będą pieniądze na dalszą modyfikację floty ochotniczych straży pożarnych. Generalnie w ratownictwie każdy nowy samochód to jest ogromna motywacja dla młodych ludzi, którzy garną się do OSP, każdy nowy samochód to jest motywacja do podnoszenia kwalifikacji. Chciałbym państwa posłów zapewnić, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie dbało o to, żeby odpowiednie środki finansowe były przekazywane na ten cel. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie ustawa ta wyjdzie z rządu, trafi do Sejmu. Tam gdzie były wątpliwości, zostały one wyjaśnione. Tak naprawdę jest to zbiór ważnych przywilejów dla środowiska, ważnych elementów dla funkcjonowania OSP, ogromne wsparcie, bo OSP buduje system bezpieczeństwa państwa, jest istotnym elementem ochrony przeciwpożarowej. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Przechodzimy do pytania drugiego.

Bardzo proszę, pytanie zadaje pani poseł Urszula Augustyn. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Pytanie skierowaliśmy także w formie interpelacji, ale odpowiedź na tę interpelację nie była dla nas satysfakcjonująca, w związku z tym chcemy dopytać, skorzystać z okazji, żeby wiedzieć na pewno. Interpelację napisaliśmy właśnie dlatego, że organizacje pożytku publicznego, które korzystają z pieniędzy, które są przekazywane przez podatników w ramach tzw. odpisu 1%, służą tym organizacjom jako źródło finansowania działalności statutowej. O tym, że organizacje pozarządowe robią bardzo dużo, wykonują bardzo dobrą robotę, nikogo przekonywać nie trzeba, natomiast pewnie należy nam się wszystkim informacja i wytłumaczenie.

A więc prawie 56 mln nie dotarło, zginęło gdzieś pomiędzy podatnikiem, który te pieniądze chciał przekazać, a organizacją pożytku publicznego, która z tych pieniędzy mogłaby skorzystać. Po pierwsze, chcielibyśmy wiedzieć, co się z tymi pieniędzmi stało. Po drugie, jaki był sposób weryfikacji? Bo czytamy w odpowiedzi na interpelację, że urzędy skarbowe zakwestionowały sposób przekazywania tych pieniędzy. Dlaczego? I wreszcie, po trzecie, czy organizacje pożytku publicznego, które były adresatami tych pieniędzy, dowiedziały się, że z jakichś przyczyn tych pieniędzy nie mają? I czy dowiedzieli się o tym ci, którzy te pieniądze przekazywali, czyli po prostu podatnicy? Bardzo proszę o odpowiedź. Zapraszam, pani minister. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli osoba fizyczna, może na zasadach i w trybie określonych w przepisach przekazać 1% podatku obliczonego zgodnie z przepisami na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Darczyńcy mają możliwość wyboru beneficjenta 1% podatku spośród organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania przedmiotowych środków, tj. figurujących w wykazie prowadzonym i publikowanym przez dyrektora Narodowego Instytutu Wolności. Zestawienie to jest ogólnodostępne, można je znaleźć chociażby na stronie instytutu.

Przepisy precyzyjnie wskazują warunki, jakie zarówno darczyńca, jak i beneficjent 1% podatku muszą spełnić, aby można było przekazać kwotę wskazaną we wnioskach na rachunki bankowe organizacji pożytku publicznego. Jednym z warunków, które muszą być spełnione, aby naczelnik urzędu skarbowego przekazał środki z 1% wskazanej przez podatnika organizacji pożytku publicznego, jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zapłata podatku musi nastąpić nie później niż w terminie 2 miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zaległość podatkowa w tym podatku nie przekracza kwoty 8,70 zł.

Pragnę poinformować, że ok. 93% podatników niestety nie wpłaciło pieniędzy, mimo że deklarowało w swoim zeznaniu, że takie pieniądze chce przekazać na organizację pożytku publicznego. Tym samym mamy 93% negatywnie zweryfikowanych wniosków o przekazanie 1%. Dotyczyło to przypadków zapłaty podatku po upływie terminu, co tym samym uniemożliwiło przekazanie 1%. Drugi przypadek: brak przekazania środków może mieć też przyczyny niezależne od tego darczyńcy, bo może wynikać z niespełnienia określonych przepisami prawa warunków właśnie przez organizacje pożytku publicznego. Np. organizacja nie podała numeru rachunku bankowego właściwego do przekazania 1% lub numer tego rachunku jest nieprawidłowy. Wtedy pieniądze wróciły. Dzieje się tak również wtedy, gdy organizacja pożytku publicznego nie figuruje lub została usunięta z wykazu Narodowego Instytutu Wolności. Odnosząc się do wskazanej kwoty prawie 56 mln zł, która nie trafiła na rachunki bankowe organizacji pożytku publicznego jako rozliczenie 1% podatku od osób fizycznych, informuję, że z danych pozyskanych od naczelników urzędów skarbowych wynika, że negatywnie zweryfikowano wnioski o przekazanie 1%, a powodem braku przekazania tych środków było właśnie niespełnienie ww. warunków, czyli albo brak zapłaty podatku w terminie, albo brak rachunku lub błędnie podany rachunek organizacji, albo usunięcie organizacji z wykazu organizacji pożytku publicznego. Weryfikacja wniosków o przekazanie 1% podatku od osób fizycznych na rzecz wybranej organizacji realizowana jest na podstawie obowiązujących i powszechnie znanych regulacji prawnych. W każdym negatywnie zweryfikowanym przypadku odstąpienie od dystrybucji wnioskowanych kwot 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. znajdowało uzasadnienie w obowiązujących przepisach prawa. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pani minister. Rozumiem, że pani poseł Urszula Augustyn z pytaniem uzupełniającym.

To po pierwsze. Po drugie, pytałam o to, czy te organizacje pozarządowe otrzymały taką informację. Może się okazać, że ktoś podał błędny numer konta, czasem to jest kwestia jednej cyfry, i może ktoś nie wie o tym, że te pieniądze mogłyby trafić na konto organizacji pożytku publicznego, ale nie trafiają ze względu na pomyłkę. A więc chcę zapytać raz jeszcze, bo pytałam o to przed chwilą, czy ktoś informuje te organizacje pozarządowe, że jest jakiś problem np. z ich adresem czy też numerem konta. Czy ktoś informuje darczyńców? Pani minister była uprzejma powiedzieć, że może ktoś tam się spóźnił, darczyńca spóźnił się z wpłatą tego podatku. Jeżeli się spóźnił, a te pieniądze chce odpisać, chce je przekazać organizacji pożytku publicznego, to czy one są przekazywane nawet po terminie, czy też nie? A jeżeli nie, to gdzie one fizycznie są? Czy ona otrzymuje informacje o stanie rzeczy? Chodzi o to, czy ktoś zdaje taki raport, żeby Rada Działalności Pożytku Publicznego mogła np. nawiązywać kontakty z organizacjami. Dziękuję, pani poseł. Bardzo proszę, pani minister, o udzielenie odpowiedzi. Wysoka Izbo! Jeszcze raz spróbuję powtórzyć.

To jest 93% przypadków. Zgodnie z przepisami prawa Urząd Skarbowy nie ma możliwości przekazania tych pieniędzy. A więc jeżeli dany podatnik rzeczywiście rozliczył się ostatecznie z fiskusem, pieniądze trafiają do budżetu państwa. Jeżeli z kolei organizacja pożytku publicznego nie zweryfikowała swojego numeru konta, nie zgłosiła go zgodnie z przepisami, to też trudno, żeby Ministerstwo Finansów informowało każdą organizację o tym, że jej rachunek bankowy jest błędny, tak?

Natomiast musimy działać jako fiskus w granicach prawa, a prawo mówi o tym, że tych pieniędzy nie możemy przekazać organizacji. Dziękuję bardzo, pani minister. Przechodzimy do kolejnego pytania. Pytanie przygotowane przez posłów Mieczysława Kasprzaka i Jana Łopatę z Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska w sprawie galopującej inflacji jest skierowane do prezesa Rady Ministrów. Bardzo proszę, pan poseł Mieczysław Kasprzak w pierwszej kolejności zadaje pytanie. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! To swoisty rekord. Węgrzy również są na tym samy poziome. Co to oznacza dla naszej gospodarki, a przede wszystkim dla Polaków?

To powoduje, że Polacy coraz mniej mogą kupić za swoją pensję, za swoje zarobki.

Z roku na rok jest o 5% środków mniej w budżetach Polaków, emerytów.

Takie są odczucia, że rządowi tak jakby zależało na tym, żeby ta inflacja była jak najwyższa, bo wtedy rząd ma większe korzyści budżetowe.

Czy rząd ma jakiś pomysł, żeby zatrzymać wzrost cen. Bo 10% to jest bardzo dużo. Dziękuję bardzo. Na pytanie odpowie, z upoważnienia prezesa Rady Ministrów, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, minister Piotr Patkowski. Bardzo proszę, panie ministrze. Wysoka Izbo! Odpowiedź na to pytanie chciałbym rozpocząć od dwóch bardzo mocnych zastrzeżeń. Po pierwsze, polityka inflacyjna w bardzo dużej mierze podpada pod Narodowy Bank Polski, Radę Polityki Pieniężnej, więc przedstawiciele rządu, a w szczególności Ministerstwa Finansów, muszą być bardzo ostrożni w wypowiadaniu się na ten temat, żeby nie posądzono ich o naruszenie niezależności tych dwóch konstytucyjnych organów. I drugie zastrzeżenie, od którego chciałbym rozpocząć i co do którego, myślę, wszyscy w tej Izbie, na tej sali się zgadzamy: niezależnie od wszelkiego rodzaju opinii czy wskaźników makroekonomicznych odczyt inflacyjny za maj - wczoraj GUS go uaktualnił, wynosi on 4,7% - jest wysoki.

Natomiast chciałbym zapewnić, że mamy świadomość, że ten majowy odczyt budzi wśród Polaków pewne obawy i niepewność. Natomiast odpowiedź na pytanie chciałbym zacząć od tego, że cel inflacyjny przyjęty przy powszechnym konsensusie ekonomistów wynosi 2,5%, z możliwymi odchyleniami zarówno w górę, jak i w dół o 1 punkt procentowy.

Pierwszy to podwyżki cen administracyjnych, na które mamy umiarkowany wpływ, bo są to ceny za usługi wodno-kanalizacyjne i ceny energii.

Druga kwestia, która wpływa na wysoki odczyt majowy, to są ceny ropy, całkowicie niezależne od rządu.

72 dolary plus słaby złoty w stosunku do dolara - to ma wpływ także na podbijanie ceny inflacji. Trzecia kwestia to odłożony popyt.

Podaż nie nadążała za popytem. Nie nadążała nie dlatego, że jest zniszczona na skutek działań wojennych, ale dlatego, że była administracyjnie zamknięta.

Czwarty bardzo istotny czynnik, który ma wpływ na inflację, to tzw. zakotwiczenie przewidywań inflacyjnych. Jest trochę tak, że im wyższe zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych, tym bardziej inflacja sama się napędza, choć statystyka ma z tym niewiele wspólnego. Dlatego to ważne - pomijając publicystyczne oceny - że jeżeli odnosimy się do makroekonomicznych wskazań, to powinniśmy być bardzo dokładni i nie używać wobec obecnej inflacji czysto technicznego, ekonomicznego terminu, jakim jest galopująca inflacja. Bo według jednolitej doktryny ekonomicznej galopująca inflacja to jest kilkanaście czy kilkadziesiąt procent i realny spadek dochodów z tytułu wynagrodzeń. Co do tego, że nie mamy inflacji w wysokości kilkunastu i kilkudziesięciu procent, nie ma wątpliwości, bo na to wskazuje GUS.

W samym sektorze przedsiębiorstw nominalny wzrost wynosi 9,9%, a realny, czyli uwzględniający inflację - 5,3%. Czyli nie mamy do czynienia ze zjawiskiem spadku realnej siły wynagrodzeń. Oczywiście dynamika osłabła, ale ciągle jest wyraźnie dodatnia.

Odpowiadając na pytania panów posłów, wyjaśnię, co jako rząd zamierzamy zrobić.

Inflacja niestety, albo stety, wymyka się czasami statystyce.

Drugi instrument - już nie behawioralny, tylko bardzo twardy - to bieżące monitorowanie, czy jako cała gospodarka nie osiągamy i nie przewyższamy luki produktowej (Dzwonek), czyli nie dostosowujemy popytu do podaży. Na szczęście - i to też wskazaliśmy w wieloletnim programie finansowym - nasz popyt maksymalny ciągle nie spełnia wszystkich możliwości podażowych polskiej gospodarki. To jest główny wskaźnik, który zapala w razie czego pomarańczową lampkę, gdy rzeczywiście inflacja wymyka się spod kontroli.

To jest główny cel, do którego Ministerstwo Finansów dąży od wielu lat i który będziemy kontynuować, jeśli chodzi o ograniczanie inflacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Zapraszam, panie pośle. Bardzo dziękuję. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie ministrze, pytamy dzisiaj o inflację, o wzrost cen, a w zasadzie o drożyznę i o to, czy ona jest galopująca, czy też nie. Wzrost cen jest bardzo wysoki, najwyższy od 20 lat, i niestety wzrasta, co sam pan przyznał.

Niestety w tej powszechnej retoryce rządowej, propagandzie wręcz o nowym ładzie, o polskim ładzie, o wzroście dochodów, jakoby wielkim - ani słowa o tym negatywnym zjawisku.

Panie Pośle! Nie oskarżam opozycji, wskazuję tylko na ten istotny czynnik behawioralny i on, chcąc nie chcąc, zawsze przy inflacji występuje. Prawidłowe zakotwiczenie celów inflacyjnych jest najskuteczniejszym sposobem walki organów państwowych, także Sejmu, z ewentualnym wzrostem inflacji. I nie możemy mówić o galopującej inflacji, kiedy doktryna inaczej ją opisuje, a mamy zupełnie inne zjawisko w polskiej gospodarce. Zgodnie z doktrynami ekonomicznymi mamy inflację na pograniczu pełzającej i stopniowej, ale nie galopującej, tak że naprawdę bym prosił, żebyśmy nie nazywali inflacji galopującą, jeśli jej nie ma, bo to nie jest inflacja galopująca i potwierdzi to każdy ekonomista. Mamy natomiast świadomość tego, że rzeczywiście ten majowy odczyt jest wysoki, tylko chciałbym wskazać na to, że mamy najprawdopodobniej ewentualnie jeszcze z odczytem czerwcowym inflacyjny pik tegoroczny. Także będziemy mieli inflację opadającą, panie pośle, i to jest kluczowa rzecz, którą chciałbym powiedzieć. Natomiast co do budownictwa. Na to znowu wpływa szereg kwestii międzynarodowych, przerwanie łańcuchów dostaw, zaburzenie podaży na światowych rynkach z tytułów obostrzeń administracyjnych, przecież one były nie tylko w Polsce, ale właściwie na całym świecie. Nie ma wyjścia.

Jeśli porównamy punktowo, o ile inflacja podskoczyła w Polsce i w Niemczech, wyjdzie nam constans i równowaga. Problem, który realnie może się pojawić - jeszcze raz to powtórzę - będzie w momencie, w którym luka produktowa spowoduje, że będziemy mieli przerost podaży nad popytem. Wtedy rzeczywiście będzie sytuacja, w której ta inflacja będzie stała i permanentna. Natomiast w tym momencie tego nie ma. Wskazaliśmy, opisaliśmy to bardzo wyraźnie w aktualizacji programu konwergencji i wskazuje na to sama Komisja Europejska. W związku z tym myślę, że to jest podstawowy wskaźnik, który na ten moment musi i powinien nas uspokoić.

Kolejne pytanie. Pytanie przygotowane przez posłów Barbarę Bartuś, Roberta Telusa i Marka Polaka z Prawa i Sprawiedliwości w sprawie uczestnictwa uczniów ze szkoły w Dobczycach w wydarzeniu politycznym Tour de Konstytucja. Pytanie skierowane jest do ministra edukacji narodowej. Pytanie zada pani poseł Barbara Bartuś. Wszystkim państwu zadającym pytanie przypominam, że aby zadać pytanie z miejsca, należy włożyć kartę do urządzenia. Bardzo proszę, pani poseł. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Dla opozycji nieważny jest młody człowiek, jego przyszłość, przyszłość narodu polskiego, przyszłość Polski. Jedynie ważna jest możliwość pewnej tuby, realizowanie własnych projektów politycznych i partyjnych oraz kształtowanie młodych ludzi według własnego pomysłu. Stąd tak zmasowany atak na polską rodzinę, na szkoły, m.in. poprzez programy seksualizujące dzieci jak Zdrovve Love w Gdańsku, a także w Łodzi, Słupsku, Warszawie.

Pamiętajmy też o tym, że to jest działanie zaplanowane, zaprogramowane i to już trwa od kilku lat. Mam tu m.in. na myśli podręcznik wydany w 2013 r. przez organizację Kampania Przeciw Homofobii. Przez tę organizację, której założycielem, pierwszym prezesem był pan Robert Biedroń. Ta książka „Lekcja równości”, która miała mówić o równości, o seksualizacji, o seksualności, była wydawana wtedy, w 2013 r., przez Związek Nauczycielstwa Polskiego jako podręcznik dla nauczycieli, jak mają postępować z dziećmi. Teraz mamy kolejny etap seksualizacji i to już na etapie nawet przedszkolaków, ponieważ na tę imprezę polityczną w Dobczycach Tour de Konstytucja zostały też zaproszone przedszkolaki. Dlatego pragnę zapytać pana ministra: Jaki jest stan faktyczny tego, co się wydarzyło w Dobczycach? I w ogóle czy ministerstwo ma wpływ na to, jak działają szkoły, na dyrektorów, na nauczycieli? Dziękuję bardzo. O udzielenie odpowiedzi na postawione pytania bardzo proszę pana ministra Tomasza Rzymkowskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Odpowiadam na zadane pytania.

Co zostało ustalone? Po pierwsze, nikt z rodziców nie wyraził zgody na udział dzieci w tym wydarzeniu. Decyzja o przyprowadzeniu dzieci na mityng polityczny została podjęta przez dyrekcję szkoły na propozycję jednej z nauczycielek, bez sprawdzenia, co to za wydarzenie i przez kogo jest organizowane. Pozwolono uczniom klas VIII i V wziąć udział w wydarzeniu o charakterze stricte politycznym. W rejestrze wyjść, obowiązkowo uzupełnianym przy wyprowadzeniu dzieci poza obręb szkoły, wpisano to wyjście dopiero w dniu przeprowadzenia kontroli, czyli już po wydarzeniu. Liczby dzieci w zapisach rejestru i w dziennikach są różne, czyli nauczyciele nie wiedzieli, ilu faktycznie uczniów mieli pod opieką. Kolejna kwestia ustalona w toku przeprowadzonej w dniu 9 czerwca kontroli.

Wysoka Izbo! Należy ponadto dodać, iż do kuratorium oświaty wpłynęły liczne skargi ze strony zaniepokojonych rodziców tychże dzieci. Stąd też czynności, które zostały podjęte przez kuratorium, były podjęte natychmiast, to znaczy następnego dnia po zdarzeniu, które miało miejsce 8 czerwca w Dobczycach. Wpłynął ponadto wniosek burmistrza Dobczyc do rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec dyrektora szkoły nr 1. Od rodziców również tego typu sygnały wpłynęły do małopolskiego kuratorium oświaty. W poniedziałek 14 czerwca dyrekcja szkoły podstawowej nr 1 zapoznała się w siedzibie kuratorium z protokołem i podpisała go. Ma w tej chwili 7 dni - ten termin zaczął biec od dnia 14 czerwca - na wniesienie poprawek, uzupełnienie bądź też sprostowanie. Wybiegając poza ten stan faktyczny, o którego przywołanie państwo prosiliście, o który zapytujecie - temu m.in. ma służyć procedowany w tej chwili przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, tak aby kurator oświaty był w stanie realnie realizować politykę oświatową państwa. Dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że my jako administracja rządowa, która odpowiada za politykę oświatową państwa, rzeczywiście możemy przeprowadzać kontrole, wizytacje, lustracje dokumentów w placówkach oświatowych, natomiast nie mamy instrumentów takich, jakie mają organy prowadzące, patrz: gminy, powiaty czy też województwa samorządowe. Ten stan rzeczy trzeba naprawić i temu ma m.in. służyć wprowadzenie mechanizmów realnego nadzoru nad kierownikami placówek oświatowych, zrównanie de facto z tymi uprawnieniami, które mają organy prowadzące wobec dyrektorów tego typu szkół, którzy nie zapewniają w naszej ocenie tych konstytucyjnych gwarancji, nomen omen, konstytucyjnych gwarancji, że to rodzice decydują o kwestiach wychowania, ale również o kwestiach światopoglądu dzieci. Natomiast te dzieci wbrew woli rodziców uczestniczyły w konkretnym mityngu politycznym, pod konkretnymi auspicjami, konkretnego środowiska politycznego. Łącznie z rzeczą absolutnie skandaliczną, to znaczy wykorzystaniem wizerunku małoletnich bez zgody rodziców w ramach akcji politycznej. Pani nie oburza to, że dzieci wykorzystane zostały do takiej hucpy politycznej? Pani poseł, naprawdę nie ma pani głosu w tej chwili. Tak, skandalem jest to, że dzieci zostały wykorzystane do hucpy politycznej. Tak, pani marszałek, to, co pani powiedziała: skandalem jest to, że dzieci zostały wykorzystane politycznie. A konstytucja mówi m.in. o promowaniu rodziny. O promowaniu rodziny, a nie homoseksualizmu i ruchów LGBT. Zdarza się właśnie tak jak w Dobczycach, że nieodpowiedzialni dyrektorzy i nauczyciele łamią prawo rodziców, rodzin, i sami decydują o kształtowaniu wychowania dzieci.

To rodzice decydują o własnych dzieciach. Powinno to być wykorzystywane. Rodzice decydują. To jest rodziców prawo i obowiązek (Dzwonek): decydowanie o wychowaniu własnego dziecka. Ja wiem, że pan mówił o dzieciach, ale tam były przedszkolaki.

Wysoka Izbo! Rzeczywiście jest tak, jak pani powiedziała. Polska konstytucja gwarantuje rodzicom wyłączność, jeśli chodzi o kształtowanie systemu wartości własnych dzieci. Szkoła polska, polski system oświaty przede wszystkim zajmuje się edukacją, ale również wspiera proces wychowawczy dzieci i młodzieży. Natomiast słowo „wspiera”, tak jak je się dobrze po polsku rozumie, oznacza, że szkoła ma wyłącznie wspierać tę wizję, którą rodzice przedstawiają. Natomiast w przywołanym przykładzie z Dobczyc widzimy sytuację skrajnie odmienną, odbiegającą od litery konstytucji, szeregu ratyfikowanych umów międzynarodowych, które gwarantują rodzicom to, że ich dzieci nie będą indoktrynowane wbrew ich woli. Tutaj mieliśmy do czynienia z sytuacją skrajnego pogwałcenia przepisów polskiej konstytucji, jeśli już o konstytucji mamy mówić. Szanowni Państwo! My, jako Ministerstwo Edukacji i Nauki, traktujemy bardzo serio kwestię ochrony polskiej rodziny. To również znajdzie swoje odzwierciedlenie w zakresie kryteriów polityki oświatowej państwa w kwestii wychowania do życia w rodzinie. Tłumaczenie, pokazywanie i wspieranie polskiej rodziny - tak, tego oczekują polscy rodzice. Polscy rodzice oczekują tego, że polska szkoła będzie edukować bardzo dobrze na bardzo wysokim światowym poziomie i będzie wspierać ich w procesie wychowawczym w coraz trudniejszych czasach. Patologią jest sytuacja, w której szkoła działa wbrew procesom wychowawczym, które wynikają z wychowania w domach. Przywołuję to i powtarzam: do Kuratorium Oświaty w Krakowie wprost tego samego dnia wpłynęły skargi ze strony zbulwersowanych rodziców, że wbrew ich woli, bez ich wiedzy ich dzieci uczestniczyły w mitingu o charakterze politycznym, podczas którego przedstawiono treści, które po pierwsze były niezgodne ze światopoglądem rodziców, a po drugie były nieadekwatne do wieku tych dzieci. To jest rzecz po prostu absolutnie skandaliczna. Bardzo się dziwię, że są środowiska polityczne w Polsce, które biorą tego typu patologiczne zachowania w obronę. Naprawdę jest to rzecz niebywała. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Przechodzimy do kolejnego pytania.

Bardzo proszę, pytanie zadaje pani poseł Marzena Okła-Drewnowicz. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Tak naprawdę to właśnie nas oburza i uważamy, że jest to skandaliczne: jak można w ogóle zmniejszać stawki na program dożywiania dzieci w szkole? Przecież od 2004 r. funkcjonuje program „Szklanka mleka” Rząd lewicowy stać było na to, żeby taki program wprowadzić. Kolejny rząd, rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u, w 2009 r. rozszerzył ten program, wprowadzając owoce w szkole. Dzieci miały możliwość zjedzenia owoców czy warzyw.

Wręcz wydaje nam się, jesteśmy przekonani, że to jest sytuacja niedopuszczalna.

Dziękuję, pani poseł. Na pytanie odpowie sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, minister Ryszard Bartosik. Bardzo proszę, panie ministrze. Szanowna Pani Marszałek! Panowie Posłowie! Ich poziom wynika wyłącznie z matematycznej kalkulacji dotyczącej zmniejszenia wartości całego koszyka dostarczanego do szkół. Dostojni państwo, sytuacja, o której mówi pani poseł, wynika z tego, że korzystamy w części z unijnego finansowania.

Jest to konsekwencją wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Wyglądało to tak, że Wielka Brytania nie wykorzystywała środków otrzymywanych z unijnego programu dla szkół.

Po brexicie takie działanie jest już niemożliwe, a budżet unijny przyznany Polsce na realizację „Programu dla szkół” zmniejszył się z tego powodu w porównaniu z bieżącym rokiem szkolnym o 12,6%. Ale jest też w tych środkach dofinansowanie z budżetu krajowego, które nie uległo zmianie i wynosi 128,1 mln zł w skali roku szkolnego.

Ich poziom wynika wyłącznie z matematycznej kalkulacji zmniejszenia wartości całego koszyka dostarczanego dla szkół. Powyższe zmiany zostały wypracowane, zaakceptowane przez przedstawicieli ministerstw oraz instytucji zaangażowanych w administrowanie „Programem dla szkół” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewnia, że realizacja „Programu dla szkół” jest monitorowana. Dostosowujemy ją również do bieżącej sytuacji. W ostatnim, trudnym roku pandemicznym dokonano kilkukrotnie zmiany przepisów krajowych w celu umożliwienia realizacji programu w czasie pandemii, tj. podczas nauki prowadzonej w trybie zdalnym.

Dziękuję bardzo, panie ministrze. Pan poseł Dariusz Joński. Bardzo proszę, panie pośle. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Pan minister przed momentem powiedział, że te obniżki wcale nie są obniżkami, jak dobrze zrozumiałem.

To jest obniżka. To niewątpliwie się nie zmienia.

Naprawdę ręce, można powiedzieć, opadają, jak się słucha tego wszystkiego. Chcę zaapelować z tego miejsca, pani marszałek, do pana ministra. Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi pana ministra Ryszarda Bartosika. Zapraszam. Wysoki Sejmie! Jeśli chodzi o kwestie związane ze zmniejszeniem finansowania z Unii Europejskiej, panie pośle, takie po prostu są fakty. Korzystaliśmy, wszystkie kraje Unii Europejskiej korzystały ze środków, które nie były wykorzystywane przez Wielką Brytanię.

Z tym nie dyskutujemy. W związku z tym dofinansowanie ze środków krajowych nie uległo zmianie. Ale rzeczywiście monitorujemy sytuację. Powiedziałem w pierwszym wystąpieniu, że w czasie trudnego roku COVID-owego zmienialiśmy te przepisy i jeżeli cokolwiek miałoby się dziać dla niekorzyść szkół i dzieci, będziemy to rozporządzenie modyfikować.

Jeżeli byłoby jakiekolwiek zagrożenie, że to wsparcie byłoby mniejsze, będziemy to rozporządzenie modyfikować, aby ono się nie zmniejszyło. Ponadto spotykamy się również z dostawcami tych środków i na ten temat będziemy rozmawiać. Jeśli będzie potrzeba, rozporządzenie będzie zmieniane.

Pytanie jest skierowane do ministra zdrowia. Pytanie zada pani poseł Anna Kwiecień. Bardzo proszę, pani poseł. Dziękuję bardzo. Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Dopiero w ostatnim roku, dosłownie w ostatnich kilku miesiącach, przypomnę tu pana prof. Zembalę, w konsekwencji protestów pań pielęgniarek i miasteczka, które było zbudowane pod ministerstwem, doszło do porozumienia i do wynegocjowania przez panie pielęgniarki tzw. dodatku zembalowego. Był to rok 2015.

Nie były.

Szanowni Państwo!

W związku z tym mam pytanie. Dziękuję bardzo, pani poseł. Na pytanie odpowie podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, minister Maciej Miłkowski. Zapraszam, panie ministrze. Dziękuję bardzo serdecznie. Pani Marszałek! Szanowni Państwo!

Od początku pierwszej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości wynagrodzenia stanowią bardzo istotny element związany z docenieniem pracowników systemu ochrony zdrowia. Pani poseł powiedziała o pierwszym porozumieniu podpisanym przez prof. Mariana Zembalę.

Przez 8 lat nie było żadnej zmiany wyceny w tym zakresie i w związku z tym dyrektorzy nie mogli podwyższać tych wynagrodzeń.

Te podwyżki były realizowane niezależnie od tego, że rząd realizował podwyżki minimalnego wynagrodzenia w całej gospodarce, które, jak pamiętamy, od 2016 r. bardzo mocno wzrastało w systemie naszego państwa.

I oczywiście odpowiednio mniej, tj. 6200 zł, 5478 zł dla lekarza, który jest na rezydenturze, a 4186 zł dla lekarza stażysty.

Dziękuję bardzo. Panie Ministrze!

Mówię to z punktu widzenia pracodawców, którzy obawiają się, czy rząd skieruje środki finansowe do placówek po to, żeby móc zrealizować tę ustawę, która weszła wczoraj w życie. Chciałabym spytać, jaką kwotę rząd musi wyasygnować z budżetu państwa na realizację ustawy, która wczoraj została przegłosowana przez Sejm, przez parlament ogólnie, i jakie to będą koszty w przyszłym roku. Dziękuję bardzo. Ponownie odpowiada podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia pan Maciej Miłkowski. Bardzo proszę, panie ministrze.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało w ubiegłym tygodniu projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów, tak jak było w latach poprzednich, gdzie to wynagrodzenie jest ustalane. System zbierania informacji na temat niezbędnych środków do realizacji tej ustawy, czyli różnicy pomiędzy aktualnym wynagrodzeniem pracowników wynagrodzeń zasadniczych a wynagrodzeniem docelowym na 1 lipca br. wraz ze wszystkimi informacjami, które dotyczą pochodnych związanych z tym wzrostem wynagrodzenia zasadniczego, czyli wszystkich dodatków, dodatków stażowych, innych dodatków, jak również dyżurów nocnych - wszystkich elementów, które są związane z podwyżką płacy zasadniczej, tak jak mówiłem, bo dotyczy to płacy zasadniczej, jak również kosztów, które są po stronie pracodawców. Te informacje zbiera Narodowy Fundusz Zdrowia. Do jutra jest termin składania uwag. Będziemy chcieli, żeby to rozporządzenie zostało opublikowane bezpośrednio po wejściu w życie nowelizacji ustawy o najniższym wynagrodzeniu w sektorze ochrony zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie te dane zbierał i później wypłacał dodatkowe świadczenia każdemu świadczeniodawcy odrębnym strumieniem finansowania przez następne okresy. Każdy podmiot dostanie dokładnie kwotę, która w całości to zabezpiecza. Te środki to 3,7 mld zł z Narodowego Funduszu Zdrowia i ok. 300 mln z budżetu sektora zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, które są przeznaczone w głównej mierze na wynagrodzenia.

Przechodzimy do kolejnego pytania. Posłowie Rajmund Miller, Monika Wielichowska, Krystyna Skowrońska, Monika Rosa, Elżbieta Gelert, Katarzyna Lubnauer, Paweł Kowal, Marta Golbik, Riad Haidar, Jerzy Hardie-Douglas i Marek Hok z Koalicji Obywatelskiej pytają w sprawie sytuacji personelu medycznego.

Panie Ministrze! Skoro jest tak dobrze, jak pan minister mówił, to dlaczego wczoraj przed Sejmem strajkowały pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, lekarze i inni? Pani poseł, pani teraz nie ma głosu. Chciałabym powiedzieć, że przez ostatnie 6 lat powiększało się zadłużenie w ochronie zdrowia. Szpitale z roku na rok zwiększały swoje zadłużenie. Samorządy musiały to pokrywać.

Czekaliśmy długo, bo prawie miesiąc, na odpowiedź, ile to będzie kosztowało. Z tej ustawy wszystkie środowiska medyczne i cała opozycja są niezadowolone. Proponowaliśmy wyższe wynagrodzenia. Mamy 100 tys. nadmiarowych zgonów. Mamy niezadowolone środowisko tych, którzy ratowali Polaków. W tym okresie zmarło 138 lekarzy, 131 pielęgniarek, 19 położnych, 16 ratowników medycznych. Proszę państwa, zarażonych było prawie 24 tys. lekarzy i ok. 59 tys. pielęgniarek, 6 tys. położnych i ok. 4 tys. ratowników medycznych. Oni zasługują na godne wynagrodzenie. A państwo wczoraj przegłosowali. Dziwię się bardzo panu ministrowi, bo nie ma ważniejszej rzeczy. Na wybory kopertowe mieliście. A zatem pytamy, kiedy państwo to zrobicie, bo przez ostatnie 6 lat wycena procedur niestety nie jest najlepsza.

Szanowny Panie Marszałku! Dziękuję, pani poseł, za pytania. To przy poprzednim pytaniu chciałem uzmysłowić. Ponieważ jest otwarta ustawa o najniższym wynagrodzeniu. Przez 8 lat się udawało, w końcu jednak personel się zdenerwował i oczekiwał od państwa jakiegokolwiek ruchu. My te elementy cały czas wyprzedzamy i cały czas nowelizacja wycen przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest realizowana, i to albo w całym zakresie, poprzez wzrost wszystkich wycen.

Oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, realizowane było porozumienie pana prof. Zembali. Później było to jeszcze dookreślone przez pana ministra Łukasza Szumowskiego. W ogóle nas interesuje głównie to, co jest zgodnie z ustawą wynagrodzeniem zasadniczym w ochronie zdrowia, i na tym się opieramy.

Na dzień dzisiejszy jeszcze mogły być stosowane dodatki wyrównawcze, ewentualnie inaczej nazwane. Jeśli chodzi o personel medyczny, to też jest dla nas bardzo istotne, aby tego personelu było więcej, bo wiemy, że w znaczącej mierze był to personel o dosyć wysokim przeciętnym wieku.

One mają zdecydowanie wyższe uprawnienia. Zrealizowaliśmy kilka nowelizacji ustaw zwiększających uprawnienia np. pielęgniarek i położnych w związku z realizacją strategii na rzecz pielęgniarstwa, która została przyjęta przez rząd.

Pozwoliło to dodatkowo, umożliwiło kształcenie większej liczby personelu i aktualnie mamy ok. 180 tys. lekarzy, to jest 14 tys. więcej, niż było 6 lat temu. Jeśli chodzi o kształcenie specjalizacyjne, również bardzo mocno staramy się, żeby każdy lekarz miał możliwość specjalizacji, w szczególności w tych specjalizacjach, które są dla nas niezbędne, priorytetowe, które są lepiej finansowane. Dodatkowe pytanie zadaje pan poseł Riad Haidar. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Druga sprawa.

A moje pytanie.

Pytanie moje jest takie: Czy teraz te szpitale będą musiały zwracać ryczałt spowodowany tym, że nie wykonały procedur? Odpowiada ponownie podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia pan minister Maciej Miłkowski. Dziękuję bardzo, także za to, że się zgadzamy, że personel jest potrzebny, należy go kształcić i należy go dobrze wynagradzać.

To są światowej i europejskiej klasy specjaliści i powinni bardzo dobrze zarabiać.

Praktycznie 100% osób otrzymuje te środki. Taka osoba podpisuje porozumienie, że chce pracować w systemie ochrony zdrowia w Polsce, nie planuje wyjeżdżać, czyli specjalizuje się po to, żeby pracować w Polsce.

To w ogóle jest sytuacja bez precedensu w ostatnich latach, że szpitale, które realizowały świadczenia w zakresie COVID-u, w szczególności w istotnym zakresie w ubiegłym roku i w tym roku, znacząco zarobiły. To był najlepszy okres tych podmiotów leczniczych, ponieważ taki był system finansowania. Płaciliśmy za świadczenia standardowe i dodatkowo za świadczenia COVID-owe.

Przechodzimy do następnego pytania. Posłowie Fryderyk Kapinos, Bolesław Piecha, Katarzyna Czochara i Tadeusz Chrzan z klubu Prawa i Sprawiedliwości w sprawie kształcenia lekarzy, pielęgniarek i techników medycznych. Pytanie zadaje pan poseł Fryderyk Kapinos. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Jednym z priorytetów rządów Zjednoczonej Prawicy jest poprawa sytuacji w systemie ochrony zdrowia.

Dotyczy to m.in. edukacji przyszłego personelu medycznego. Dzięki temu w ostatnich latach stopniowo rośnie liczba lekarzy i pielęgniarek. Sukcesywnie rząd Zjednoczonej Prawicy podnosi także wynagrodzenia personelu medycznego. Wszyscy pracownicy medycznie powinni być godnie wynagradzani za swoją ciężką pracę.

Problem z liczbą personelu medycznego rząd odziedziczył po poprzednikach. Niestety, ich rządy i brak realnych działań doprowadziły do zmniejszenia liczby personelu medycznego. Rząd Zjednoczonej Prawicy nie jest obojętny w tej sprawie. Za rządów koalicji PO-PSL na koniec 2010 r. liczba lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód wynosiła 154 536 osób. Dzięki staraniom rządu Zjednoczonej Prawicy ta liczba systematycznie wzrasta. Na koniec 2020 r. mieliśmy 181 151 lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód. To wzrost liczby personelu medycznego o ponad 26 tys.

Chciałbym zadać pytanie.

Bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku! Dziękuję bardzo serdecznie. Kolejne pytanie dotyczące kadr w ochronie zdrowia i kadr, które odziedziczyliśmy.

Jeśli chodzi o personel lekarski, to pierwsza, podstawowa rzecz, Ministerstwo Zdrowia poprzez zwiększenie limitów na studia, poprzez zwiększenie liczby miejsc udzielania świadczeń, miejsc kształcenia personelu medycznego poprzez budowę nowych uczelni medycznych zwiększyło możliwości przyjęć na kierunek lekarski o 2 tys. miejsc, tj. o ok. 1/4.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w której planujemy uruchomienie kredytu na studia, który będzie realizowany na rzecz kształcenia, który będzie pod określonymi warunkami umarzany tym osobom, które będą pracowały w Polsce. Dodatkowo żeby ten zasób uczelniany powiększyć i polepszyć, bardzo wiele środków było przeznaczanych na wyposażenie, na zwiększenie możliwości kształcenia personelu medycznego i obecnie w Krajowym Planie Odbudowy na lata przyszłe zostały zabezpieczone środki w wysokości 700 mln euro dla uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych dwóch głównych grup zawodowych, czyli pielęgniarek i lekarzy.

To są 22 specjalności.

Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Liczba szkół posiadających akredytację Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie studium na kierunku pielęgniarstwa na

Szkolenie rezydenckie w tym roku rozpocznie aż 900 lekarzy, a w 2015 r. rozpoczęło je 300 lekarzy. I mam dodatkowe pytanie: Jakie działania będzie podejmowało Ministerstwo Zdrowia w najbliższych latach, aby zwiększyć liczbę wykwalifikowanych nie tylko lekarzy - to już pan minister powiedział - lecz także pielęgniarek i ratowników medycznych? Dziękuję bardzo. Pan minister Maciej Miłkowski.

Zwiększamy te możliwości.

Mogą również samodzielnie realizować porady ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Ustaliliśmy, że pielęgniarki i położne bez dodatkowych kursów mogą kwalifikować do szczepień przeciwko COVID-19 i je wykonywać.

To też jest istotne.

Przechodzimy do następnego pytania.

Panie Ministrze! Cieszy tempo i skala budowy dróg w całej Polsce za rządów Prawa i Sprawiedliwości, w tym budowa dróg ekspresowych. One powinny tworzyć, tak jak zresztą wszędzie, spójny i funkcjonalny układ komunikacyjny. Tak by było, gdyby ten plan budowy dróg ekspresowych w tym rejonie Polski nie został dotknięty pewną wadą, którą pan minister zna, bo nieraz o tym rozmawialiśmy. Ta wada polega na tym, że od 2009 r., kiedy zmieniono przebieg dróg ekspresowych w województwie podlaskim - to było za czasów rządów PO-PSL - odcinek bardzo ważny, uczęszczany, obciążony ruchem tranzytowym, ruchem ciężarowym, Białystok - Augustów, został wyłączony z tej sieci dróg ekspresowych. Drogi trzeba budować tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Pan minister Andrzej Adamczyk zawsze to twierdzi. To bardzo mądre, ważne zdanie. I właśnie niezrozumiała jest sytuacja, która polega na tym, że ta sprawa nie została uregulowana i przywrócona od czasów rządów PO-PSL.

w imieniu nie tylko własnym, ale też wszystkich parlamentarzystów województwa podlaskiego, licznych mieszkańców, którzy. Odpowiada sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury pan Rafał Weber. Proszę, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Rozwój sieci drogowej w każdym regionie Polski jest priorytetem rządu Prawa i Sprawiedliwości, priorytetem Ministerstwa Infrastruktury. Nowoczesna infrastruktura zapewnia bezpieczeństwo, płynność ruchu, wygodę i komfort jazdy. Tworząc spójną sieć, zwiększamy dostępność transportową, tak ważną w kontekście rozwoju społecznego i gospodarczego. Sprawne rozwiązania komunikacyjne są czymś, co w ewidentny sposób wpływa na podniesienie statusu i wartości danego regionu. Bez dróg szybkiego ruchu bądź bez niwelacji wąskich gardeł przelotowych ciężko mówić nie tylko o odpowiednich warunkach do właściwego komunikowania się społeczeństwa, ale też o odpowiednich warunkach do prowadzenia biznesu. I właśnie przez ten pryzmat Ministerstwo Infrastruktury patrzy na inwestycje drogowe. Widzimy w nich warunek sine qua non szans rozwojowych we wszystkich aspektach. Przechodząc do przedmiotu pytania pana posła Jarosława Zielińskiego czy grupy posłów, pytania dotyczącego rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Białystok - Augustów, chcę potwierdzić zamiary Ministerstwa Infrastruktury podniesienia jakości tej drogi nawet do parametrów, które w pewnym stopniu odpowiadają drogom ekspresowym.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku analizuje tę kwestię i sześćdziesiątkę jedynkę oraz S19 połączymy właśnie tym korytarzem poprzez rozbudowę czy nowy ciąg równoległy do drogi krajowej nr 8 albo korytarzem między Knyszynem a Ełkiem. W tej chwili dwa warianty wchodzą w grę. Efekty tych prac poznamy w IV kwartale tego roku.

Tak jak mówię, pod koniec tego roku, po analizach, które w tej chwili są prowadzone, rozstrzygnie się, który z tych wariantów będzie realizowany. Natomiast żeby nie czekać tylko i wyłącznie na te kwestie, wprowadzimy inwestycje polegające na budowie obwodnic w ciągu drogi krajowej nr 8. Dzięki rządowemu programowi budowy 100 obwodnic obwodnica Sztabina, czyli tej miejscowości, o której wspominał pan poseł, a także obwodnica Suchowoli oraz Białobrzegów - te inwestycje znalazły się w rządowym programie budowy 100 obwodnic. Są one na liście podstawowej, mają zabezpieczone środki finansowe, co ważne, i są realizowane. W przypadku obwodnic Suchowoli i Sztabina w grudniu poprzedniego roku ogłoszone zostały przetargi na wybór wykonawców, zaś w przypadku obwodnicy Białobrzegów ten przetarg zostanie ogłoszony w przyszłym roku. W tej chwili jest opracowywana koncepcja programowa. Umowa na wykonanie obwodnicy Suchowoli została zawarta 14 maja br., natomiast 28 maja br. została podpisana umowa na obwodnicę Sztabina. I chcę podkreślić, że to są umowy wykonawcze. Pozostały więc kwestie projektowe, później uzyskanie pozwoleń budowlanych i wejście na plac budowy.

Dzięki budowie tych obwodnic nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców tego regionu. Nastąpi odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości drogi krajowej nr 8 między Białymstokiem a Augustowem na odcinku ok. 25 km. W przypadku odcinków międzyobwodnicowych na ósemce należy wskazać, że do chwili obecnej zostały uzyskane ostateczne decyzje środowiskowe, co jest bardzo ważne, bo praca nad decyzjami środowiskowymi jest bardzo czasochłonna i coraz trudniejsza.

Apeluję o zmianę perspektywy myślenia.

Dlaczego resort się upiera, żeby nie przywrócić tego pierwotnego, dobrego planu? Naprawdę wszystkie argumenty świadczą za tym, żeby tak było. Panie Ministrze! Ogromna prośba o zmianę perspektywy patrzenia na tę sprawę. Odpowiada ponownie sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury pan Rafał Weber. Szanowni Państwo!

Ona jest w realizacji na wszystkich odcinkach.

Po zakończeniu tej inwestycji to ona przejmie niemalże cały ruch tranzytowy biegnący w kierunku Litwy i dalej, do państw nadbałtyckich.

Natomiast jeżeli chodzi o rozbudowę DK8, to w jednym z wariantów idziemy dalej, niż pan poseł wnosi.

Tak że być może, podkreślam: być może - a wyjdzie to z analiz środowiskowych, technicznych, ekonomicznych i oczywiście społecznych - pójdziemy dalej, niż pan poseł ma na myśli, dalej niż pan poseł to artykułuje.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i bardzo wysoka kwota na województwo podlaskie. Tylko jeden powiat. Tak że mówienie o tym, że Ministerstwo Infrastruktury nie realizuje potrzeb komunikacyjnych w woj. podlaskim jest. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do kolejnego pytania. Jako pierwsza pytanie zada pani poseł Teresa Pamuła. Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! Inwestycje drogowe mają kluczowe znaczenie dla rozwoju nie tylko komunikacyjnego czy transportowego, ale i kompleksowego rozwoju Rzeczypospolitej. Spójna sieć dróg bezpiecznych, wygodnych i komfortowych to klucz do podniesienia potencjału gospodarczego poszczególnych regionów Polski. Obecnie Ministerstwo Infrastruktury realizuje zadania drogowe m.in. poprzez „Program budowy dróg krajowych” z perspektywą do 2025 r. W ramach tego programu sieć dróg szybkiego ruchu jest rozbudowywana o tysiące kilometrów. W każdym, podkreślam: w każdym, regionie Polski prowadzone są inwestycje. Strategiczną dla Podkarpacia inwestycją drogową jest Via Carpatia. Połączenie na osi Północ - Południe dla mojego województwa jest szansą na usprawnienie komunikacyjne i dużo lepszy kontakt nie tylko z innymi regionami naszego kraju, ale też z państwami sąsiednimi. Via Carpatia to szlak, który łączy kraje nadbałtyckie z państwami na południu Europy. Międzynarodowy charakter tej drogi sprawia, że przez Polskę będzie przebiegać jeden z głównych korytarzy Starego Kontynentu. To, że ta inwestycja jest prowadzona, wynika ze strategii rozwojowej rządu Prawa i Sprawiedliwości. Niwelacja wykluczenia komunikacyjnego regionów mniej rozwiniętych jest celem działania rządu i Ministerstwa Infrastruktury. Właśnie poprzez „Program budowy dróg krajowych” nadrabiamy zaległości inwestycyjne. Gdyby nie obecne decyzje rządu, wiele z inwestycji po prostu nie byłoby realizowanych, a Via Carpatia jest tego najlepszym przykładem. Rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego nie widział potrzeby zabezpieczenia finansowego dla tej inwestycji.

Panie Ministrze! Proszę o informację, [[Dzwonek]] jak obecnie wygląda realizacja „Programu budowy dróg krajowych” Ile zadań jest w fazie wykonawczej, a ile w pracach przygotowawczych?

Panie Marszałku! Pani Poseł! Szanowni Państwo!

Dzięki staraniom ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka w ciągu ostatnich 5 lat limit tego programu podnoszony był kilkukrotnie, a podniesienie limitu to nowe inwestycje, które mają zabezpieczenie finansowe i mogą być realizowane. Pierwotna wartość programu to 107 mld zł, to jest ta wartość z końca 2015 r., a obecna wartość to 164 mld zł, czyli o 57 mld zł więcej. I to jest miara autentycznej skuteczności ministra Andrzeja Adamczyka, ale też całego rządu Prawa i Sprawiedliwości, teraz pana premiera Mateusza Morawieckiego, a wcześniej pani premier Beaty Szydło, bo limit zwiększany był uchwałą rządu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że infrastruktura drogowa jest ważnym elementem, takim niezbędnym czynnikiem prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki całej Rzeczypospolitej. Nowoczesna i spójna sieć drogowa jest jednym z celów, do jakich Polska dąży w ostatnich latach.

Łącznie, biorąc pod uwagę same kilometry, jest to prawie 80% planowanej długości nowych dróg szybkiego ruchu w Polsce.

To jest najlepszy dowód na to, że potrafimy skutecznie i efektywnie prowadzić prace inwestycyjne, pomimo trudnych okoliczności, np. pandemicznych, które przecież od ponad roku występują. Co ważne, szanowni państwo, inwestycje drogowe prowadzone są w każdym regionie naszego kraju. Podkreślam: w każdym. W każdym województwie.

Inwestycje w drogi szybkiego ruchu prowadzone są w każdym regionie, we wszystkich 16 województwach naszego kraju. Natomiast odnosząc się do Via Carpatii - tak, faktycznie, to jest jedna z kluczowych inwestycji, które są realizowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Oczywiście rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u miał inne plany, nie widział sensu w budowie tej drogi. nawet przedstawiciele Platformy Obywatelskiej ostro protestowali przeciwko. w Parlamencie Europejskim w 2014 r. Ale my jako Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie od momentu przejęcia odpowiedzialności za polskie sprawy realizujmy Via Carpatię. Przeznaczamy na jej budowę blisko 30 mld zł. Znaczna część tych środków finansowych została zapewniona w programie budowy dróg krajowych w roku 2017. Później, przy kolejnych nowelizacjach tego programu, te środki były sukcesywnie powiększane, sukcesywnie poszerzane. Tak że tak wygląda obraz inwestycji drogowych, inwestycji polegających na budowie dróg szybkiego ruchu w ramach programu budowy dróg krajowych. Konsekwentnie, z wielką determinacją, pomimo trudności pandemicznych realizujemy zamierzone cele i mamy nadzieję, że obraz rzeczywistości drogowej w Polsce będzie zmieniał się nadal bardzo szybko. Bardzo proszę. Dziękuję, panie ministrze, za udzielone informacje. Zależy nam bardzo na tym, aby nowoczesna infrastruktura funkcjonowała jak najszybciej, bo ona ma całościowy wpływ na rozwój Polski. Chciałabym usłyszeć jeszcze, jaki jest stan zaawansowania realizacji Via Carpatii. Jak rysuje się wykonanie tej inwestycji na południe od Rzeszowa do granicy w Barwinku? Ta droga jest niezbędna od strony rozwoju społecznego i dlatego zależy nam na jej wykonaniu. Ale wiemy doskonale, że nie chodzi tylko o Podkarpacie, choć zadaję pytania dotyczące odcinków m.in. tam budowanych, bo to ma znaczenie międzynarodowe i to bardzo ważna droga dla naszego kraju.

Korzystając też z obecności na sali byłego ministra infrastruktury, który tutaj mówił o Via Carpatii i o tym, że chciał ten projekt realizować, powiem, jak został ten projekt zrealizowany właśnie przez Platformę Obywatelską na odcinku podkarpackim Jasionka - Sokołów Małopolski.

Ale ten błąd naprawiamy. Ten błąd naprawiamy. polegający na dobudowie kolejnego pasa na tym odcinku Via Carpatii. Wracając do pytania pani poseł - pierwsze odcinki Via Carpatii między Rzeszowem a Lublinem będą oddawane do użytkowania już w tym roku. Ba, nawet jeden w ostatni poniedziałek został oddany w ramach czasowej organizacji ruchu. Za rok stolice województw lubelskiego i podkarpackiego będą połączone drogą szybkiego ruchu, właśnie Via Carpatią. Jeżeli mówimy o odcinkach na południe od Rzeszowa, to ten z bardzo długim tunelem między Rzeszowem Południe a Babicą jest już projektowany.

Ale naprawdę warto, to się opłaci, ta droga zaprocentuje. Pozostałe dwie umowy zostaną podpisane w najbliższym czasie, a z biegiem tego roku będą ogłaszane ostatnie bodajże trzy przetargi na budowę tych odcinków między Rzeszowem a granicą państwa ze Słowacją. Sześć umów na realizację zostało podpisanych w województwie podlaskim. Kolejne przetargi są przygotowywane i będą sukcesywnie ogłaszane.

Nie pozostaje nam nic innego, jak zgodnie z deklaracjami, zgodnie z obietnicami realizować tę inwestycję, ale - tak jak powiedziałem wcześniej - też szereg innych inwestycji, drogę ekspresową S14 w województwie łódzkim (Dzwonek), również po to, aby polepszać infrastrukturę drogową w naszym kraju. Przechodzimy do następnego pytania. Posłowie Krzysztof Gawkowski, Robert Obaz, Magdalena Biejat, Anita Kucharska-Dziedzic, Marek Rutka, Joanna Senyszyn, Przemysław Koperski, Dariusz Wieczorek, Monika Falej, Paulina Matysiak, Katarzyna Kotula, Robert Kwiatkowski, Karolina Pawliczak, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Paweł Krutul, Lewica, kierują pytanie w sprawie przebiegu negocjacji ze stroną czeską przed wydaniem przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazu natychmiastowego wstrzymania wydobycia węgla oraz wstrzymania prac w kopalni Turów i po jego wydaniu - do prezesa Rady Ministrów. Bardzo proszę, panie pośle. Wysoka Izbo! Pan jest tak naprawdę twarzą tego, co się dzieje w tych negocjacjach. Pomaga panu pan minister Sasin, ale on ma doświadczenie tylko w organizacji wyborów. Traktujecie mieszkańców Bogatyni, powiatów: zgorzeleckiego, lubańskiego, bolesławieckiego jak pionki na szachownicy, które przestawiacie w zależności od potrzeb politycznych. Najpierw przy protestach Czechów od roku 2016 kompletnie nic nie robiliście, a na konsultacje społeczne z mieszkańcami pogranicza czeskiego zaprosiliście tłumacza, który nie znał języka technicznego.

Teraz pojawiają się sprzeczne informacje, że kopalnia, owszem, będzie funkcjonować, ale być może nie tak długo, jak zakłada to przedłużona koncesja na wydobycie węgla. Tylko znowu pojawia się pytanie: Co z mieszkańcami, co z miejscami pracy? Dlatego też, panie premierze, chciałbym zapytać: Jak konkretnie przebiegały negocjacje ze stroną czeską, zarówno do czasu ogłoszenia postanowienia TSUE nakazującego wstrzymanie prac w kopalni, jak i tuż po jego ogłoszeniu? Ile odbyło się spotkań negocjacyjnych, w jakich terminach i w jakim składzie? Co konkretnie jest przedmiotem negocjacji i na jakim etapie dzisiaj znajduje się przygotowanie porozumienia oraz na kiedy planowane jest jego podpisanie? Biorąc pod uwagę konsekwencje zamknięcia kopalni, a w perspektywie także wygaszanie elektrowni, w jaki sposób pański rząd zamierza zapewnić regionowi Bogatyni i tysiącom jego mieszkańców bezpieczeństwo społeczno-gospodarcze? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.

Wysoka Izbo! Postaram się państwu w miarę obszernie przekazać informacje na temat tego, co zrobił rząd, jak wygląda sytuacja w Bogatyni i kopalni Turów, opierając się na faktach, na tym, co zostało spisane. Wydaje mi się, że jest celowe, abyśmy w tej chwili państwu to przekazali. Na wstępie chciałbym państwu powiedzieć, że rząd Rzeczypospolitej Polskiej przykłada najwyższą wagę do znalezienia możliwości polubownego rozwiązania i zakończenia sporu z Republiką Czeską odnośnie do potencjalnych skutków działalności kopalni Turów. Na przestrzeni ostatnich lat utrzymywane były stałe kontakty na poziomie roboczym pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w zakresie współpracy dotyczącej transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko dla obszaru kopalni Turów. Odbywały się też regularne spotkania na poziomie ministerialnym.

Pragnę państwu przypomnieć, że kopalnia funkcjonuje od 100 lat.

W połowie 2019 r. nastąpiła mocna intensyfikacja podnoszenia przez stronę czeską problemu działalności kopalni Turów.

W marcu 2020 r. czeski wiceminister środowiska Vladislav Smrz wprost przyznał, że sprawa jest polityczna i związana z wyborami regionalnymi.

Republika Czeska skierowała do Komisji Europejskiej skargę na domniemane naruszenie prawa europejskiego przez Rzeczpospolitą Polską w związku z przedłużeniem i rozszerzeniem koncesji na działalność wydobywczą w Turowie. Kolejno.

30 października Rzeczpospolita Polska sporządziła uwagi na piśmie i przekazała je odnośnie do skargi Republiki Czeskiej. Kolejno przedstawiciele Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyli w wysłuchaniu przez Komisję Europejską w dniu 13 listopada, które odbyło się online, podczas którego zostały przedstawione argumenty strony polskiej. To była długa dyskusja i takich spotkań, które poprzedzały to spotkanie 13 listopada, było więcej.

Te roszczenia opiewały na ponad, mówiąc otwarcie, 60 mln euro.

Myślę, że państwo jesteście przekonani, że my z naszej strony zrobiliśmy to, co do nas należy, i właściwie zrobiliśmy. Zaraz będziemy na ten temat rozmawiać. Szanowni Państwo! To jest ten dialog, który był prowadzony od 2019 r. Zaproponowaliśmy nasze rozwiązania. Częściowo wpasowały się one zarówno w zainteresowanie strony czeskiej, jak również były uzgodnione oczekiwania po stronie czeskiej. Dochodziło do dyskusji na temat ekranu przeciwfiltracyjnego, budowy specjalnej kurtyny ziemno-leśnej czy ziemno-drzewnej, która będzie zasłaniała od pyłu, hałasu i będzie stanowiła taką osłonę wizualną przed kopalnią od strony czeskiej.

Oczywiście pośrednio ma, bo lej depresyjny jest i powstaje, niemniej jednak nie chcą uznać naszych argumentów w tym zakresie, że na terenie Czech, czyli w strefie przygranicznej, bezpośrednio występuje duża żwirownia właśnie w obszarze ujęcia wody Uhelná, która jest dla nas konfliktowym problemem, gdzie lej depresyjny, który powstaje, pobiera tę wodę z ujęcia wody Uhelná. W związku z tym mamy taki problem: oni nie dostarczają nam informacji, danych, a my dane, które posiadamy, pokazujemy, zaś oni nie chcą ich tak naprawdę zaakceptować.

I to jest ta historia, którą w skrócie chciałem przedstawić. Oczywiście jesteśmy na takim etapie, na jakim jesteśmy. Uznajemy tutaj rezultat Komisji Europejskiej, wynik oceny.

To wiecie. To wszystko wiecie państwo, tak?

Bardzo proszę, pytanie dodatkowe, pan poseł Robert Obaz. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Najważniejszą rzeczą. Liczę na to, że na te wszystkie pytania otrzymam odpowiedź na piśmie, w imieniu wszystkich posłów, którzy się pod tym podpisali. Ale, panie ministrze, co dalej z transformacją tego regionu?

Dziękuję bardzo. Panie ministrze, bardzo proszę jeszcze raz, jeżeli pan zechce, ale już tak bardzo skrótowo. Bardzo krótko. Szanowny Panie Pośle!

Nasiliły się przed wyborami samorządowymi i w tej chwili przed wyborami, jest to sprawa bardzo wyraźnie polityczna. Jeszcze co do petycji mieszkańców - ci sami mieszkańcy również napisali petycję, że żądają utrzymania kopalni. Ale piszą o utrzymaniu kopalni, tak? O prowadzeniu działalności eksploatacyjnej. Potwierdzam, ekran jest. Nawet widziałem pewne protokoły odbioru, które są już z marca, częściowe oczywiście. Wykonanych jest 200, z tego, co pamiętam, 200 otworów iniekcyjnych - też na dzień dzisiejszy - tyle, ile jest planowanych. Natomiast drugą kwestią, jeśli chodzi o ekran, jest to, że jeśli ten ekran nie będzie zdawał egzaminu na tyle, na ile zostało to założone - bo to jest zawsze założenie projektowe - to PGE jest zainteresowane, żeby w trybie szybkim, pilnym rozszerzyć ekran i go pogłębić. Dziękuję bardzo, panie ministrze. To pytanie kończy rozpatrywanie tego punktu porządku dziennego. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 3. porządku dziennego: Informacja bieżąca. Przypominam, że na obecnym posiedzeniu Sejmu zostanie rozpatrzona informacja w sprawie bezpieczeństwa energetycznego Polski (kopalnia Turów, zielona transformacja, Baltic Pipe, fotowoltaika, Elektrownia Bełchatów), o której przedstawienie wnosił Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni. Przypominam również, że przedstawienie uzasadnienia wniosku przez posła przedstawiciela wnioskodawców nie może trwać dłużej niż 5 minut, a udzielenie odpowiedzi przez przedstawiciela Rady Ministrów - dłużej niż 10 minut. Wystąpienia posłów w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż 2 minuty. Na zakończenie dyskusji głos zabierają kolejno przedstawiciel wnioskodawców oraz przedstawiciel Rady Ministrów. Wystąpienie przedstawiciela wnioskodawców nie może trwać dłużej niż 5 minut, a wystąpienie przedstawiciela Rady Ministrów - dłużej niż 10 minut. Marszałek Sejmu może wyrazić zgodę na wydłużenie wystąpienia przedstawiciela Rady Ministrów. Czas przeznaczony na rozpatrzenie punktu: Informacja bieżąca nie może być dłuższy niż 90 minut. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela wnioskodawców pana posła Tomasza Piotra Nowaka. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Informacja bieżąca w sprawie bezpieczeństwa energetycznego Polski z uwzględnieniem kopalni Turów, zielonej transformacji, Baltic Pipe, fotowoltaiki, Elektrowni Bełchatów. Gdzie jesteśmy w sprawie bezpieczeństwa energetycznego? Przez całą poprzednią kadencję i część obecnej rząd PiS śnił sen o węglowej potędze, tracąc lata na konieczność zmian transformacyjnych, występując przeciwko OZE, np. ustawa 10H, czy nie rozbudowując sieci tak, aby mogły przyjąć rosnącą produkcję prosumencką np. w fotowoltaice. Kolejne wersje polityki energetycznej Polski nie kreśliły zmian w potrzebnej skali. Państwo nadal blokuje rozproszoną obywatelską energetykę, wspierając niewydolne koncerny energetyczne, bowiem nadal są długotrwałe procedury w zakresie rozwoju OZE, brakuje jasnych reguł postępowania organów publicznych, np. RDOŚ. Rząd robi krok do przodu, jak np. z finansowaniem programu „Mój prąd”, a później się cofa, wprowadzając zdecydowanie gorsze rozwiązania dla fotowoltaiki i hamując jej rozwój. Nadal nie ma ustawy wprowadzającej nowy rodzaj prosumentów, np. prosumentów zbiorowych czy prosumentów wirtualnych.

To jest wynik błędnej polityki rządu, tak jak pozostawienie np. PGE i kopalni Turów samych sobie. Co prawda przed chwilą słyszeliśmy o całym harmonogramie rozmów ze stroną czeską, ale liczy się finał, a finał to krach dyplomacji biznesowej.

To jest szokujące, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie przyjął obiektywnie argumentów, które powinny spowodować to, że nie zapadnie taki wyrok. Pytanie, kto prowadził te negocjacje i jakie były argumenty. W specjalnym stanowisku podczas posiedzenia komisji zażądaliśmy także od premiera, żeby w sytuacji kryzysowej, w jakiej jesteśmy, skutecznie przeprowadził negocjacje zabezpieczające funkcjonowanie kopalni Turów. Posłowie PiS byli temu przeciwni. Nie chcą, żeby premier zaangażował się w te negocjacje. Dlaczego? Czy też uważają, że problem Turowa rozwiąże się sam, może przez ministra Sasina, zobaczymy. Do tego nakłada się awaria w Bełchatowie i konieczność odpowiedzi na pytanie, co dalej z tą największą elektrownią. Co z atomem w Bełchatowie, w Pątnowie? Nadal nie wiemy, czy Polska przyjmie neutralność klimatyczną w 2050 r. i nie wiemy, czy będzie miało wobec nas zastosowanie warunkowości ograniczającej Fundusz Sprawiedliwej Transformacji o 50%. Brakuje dokumentu strategicznego transformacji polskiej energetyki i przemysłu - środki z KPO, funduszu modernizacyjnego, wpływy ze sprzedaży uprawnień do emisji

Co z notyfikacją w Unii Europejskiej? Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska pana ministra Piotra Dziadzię. Bardzo proszę. Szanowni Państwo! Jeszcze pozwolę sobie uzupełnić te informacje, których nie zdążyłem uzupełnić, dlatego że, jak państwo widzicie, 5 minut na przedstawienie krótkiej informacji w zakresie Turowa nie wystarcza, nawet 10 minut nie wystarcza. Szanowni Państwo!

Polityka energetyczna jest planem działalności na rzecz unowocześnienia i modernizacji sektora energii oraz przeprowadzenia przekształceń w sektorze energii w sposób odpowiedzialny, efektywny, skuteczny, z zagwarantowaniem bezpieczeństwa energetycznego. W strategii wymienione zostały inwestycje mające na celu zwiększenie udziału energii z niskoemisyjnych źródeł energii oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazów cieplarnianych. To mówi o komplementarności tej polityki. Jednym z największych wyzwań, z którymi musimy się zmierzyć, będzie zagwarantowanie realizacji celów polityki klimatyczno-energetycznej w toku sprawiedliwej transformacji, przyczyniające się do poprawy jakości powietrza i stanu środowiska. Dążymy do tego, aby zmiany miały charakter partycypacyjny, czyli były prowadzone lokalnie, z uwzględnieniem aktywnej roli odbiorców końcowych. Co wymaga podkreślenia w tym kontekście? Po pierwsze, podstawą jest tutaj, i będzie, determinacja w zakresie bezpieczeństwa energetycznego poprzez pokrycie zapotrzebowania na moc własnymi zasobami wytwórczymi. Dokument ten przewiduje oddanie do eksploatacji w Polsce elektrowni jądrowej o łącznej mocy zainstalowanej pomiędzy 6 a 9 GW. Pierwszy blok jądrowy będzie oddany do eksploatacji do roku 2033. Technologia jądrowa i jej znaczenie, państwo to wiecie, pominę to i nie będę uzasadniał, dlaczego jest ona taka istotna dla bezpieczeństwa energetycznego. Do czasu zapewnienia stabilnej podstawy pracy systemu elektroenergetycznego, czyli do czasu wybudowania elektrowni, powstania energetyki jądrowej, konieczne jest zapewnienie dyspozycyjnych i sterowalnych mocy w celu zabezpieczenia systemu. Głównym instrumentem, który ma zapewnić wprowadzenie do systemu nowych jednostek, jest rynek mocy. W tym miejscu pragnę zasygnalizować, że Rada Ministrów wczoraj przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rynku mocy, którego celem jest zwiększenie efektywności tego instrumentu.

Efekt zadziałania rezerwy pierwotnej w systemie Europy kontynentalnej spowodował natychmiastowy dopływ mocy do krajowego systemu elektroenergetycznego, uzupełniając ubytek mocy.

System zadziałał prawidłowo, co oznacza, że nie było zagrożenia w zakresie odłączenia odbiorców. W tym miejscu należy odnieść się do konsekwencji postanowienia tymczasowego wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości, dotyczącego natychmiastowego wstrzymania wydobycia w Kopalni Węgla Brunatnego Turów, o czym chcę państwu powiedzieć.

Polska polityka energetyczna wskazuje w tym zakresie na główną rolę gazu ziemnego jako paliwa przejściowego. PEP 2040 wyznacza ramy zarówno inwestycji w źródła wytwórcze, jak i dywersyfikacji dostaw oraz rozbudowy infrastruktury sieci gazowej - stanowi to trzeci cel szczegółowy polityki energetycznej. W ramach tego celu projektem strategicznym jest budowa Baltic Pipe.

Jesteśmy w tym zakresie w stałym kontakcie ze stroną duńską, z władzami duńskimi, inwestorami, którzy stale nas informują o sytuacji.

Widzimy tutaj dość dużą wolę i determinację ze strony naszych duńskich partnerów, ażeby zakończyć tę inwestycję, i trzeba im za to podziękować.

Baltic Pipe jest częścią polityki dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski, skutecznie realizowaną od 2015 r.

W ramach transformacji energetycznej wzrastać będzie udział OZE przy jednoczesnym niezbędnym rozwoju elastycznych mocy rezerwowych, infrastruktury sieciowej oraz magazynowania energii.

Zakłada się, że produkcja z morskich farm wiatrowych będzie miała większy udział w produkcji energii elektrycznej wytwarzanej z OZE.

Istotnym atutem OZE jest możliwość wykorzystania potencjału lokalnego, w tym słabiej rozwiniętych regionów i obszarów wiejskich. Energetyka ta powinna jednak służyć wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycznego, uzupełniać generację źródeł centralnych i przenosić utrzymanie samowystarczalności energetycznej na poziom lokalny - takie są założenia. Konsumenci, odbiorcy aktywni, w tym prosumenci, spółdzielnie, społeczności energetyczne i klastry odgrywają główną rolę w dążeniu do osiągnięcia elastyczności niezbędnej do dostosowania systemu energii elektrycznej opartego na energetyce rozproszonej. Bez elastyczności zapewnianej przez odbiorów energii transformacja sektora energii wydaje się niemożliwa. co związane jest przede wszystkim z rozwojem takich programów, jak „Mój prąd”

Dlatego właśnie zostały podjęte takie działania. Zaproponowaliśmy m.in. innowacyjne rozwiązania niezbędne do poprawy funkcjonowania rynku energii i ten nowy system, który został zaproponowany, jest zgodny i wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i z prawa europejskiego. Nowy system prosumencki zachowa przy tym podstawowy cel. Prosument będzie posiadał możliwość obniżenia rachunków za energię elektryczną.

Dziękuję bardzo. Zamykam listę. Jako pierwszy pan poseł Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma pana posła. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciałem, po pierwsze, wyrazić uznanie - a z drugiej strony zdziwienie - dla pana Tomasza Nowaka, że w tak krótkim czasie zawarł tyle nieprawd, przeinaczeń, kłamstw i w gruncie rzeczy krytyki, choć za krytykę nie mogę go zganić, bo Platforma, a właściwie opozycja niczego innego nie potrafi poza krytyką. Szanowni państwo, mam tylko 2 minuty. Jeden aspekt, który tutaj pan poseł poruszył, jest taki, że posłowie byli przeciwni szybkim, skutecznym negocjacjom z udziałem premiera. Otóż podczas posiedzenia komisji, bo mieliśmy wiele posiedzeń komisji poświęconych energetyce, dwa na temat Turowa, państwo w gruncie rzeczy żądaliście, żeby polski rząd zawarł szybko porozumienie na warunkach czeskich, niezależnie od tego, czy Czesi mają rację, czy nie mają racji. Cała ta debata pokazywała, że Czesi próbują od nas przy okazji wyciągnąć jak największe pieniądze. Mamy w Polsce opozycję, która w gruncie rzeczy staje po stronie Czech i jeszcze popędza rząd, żeby jak najszybciej zawarł to porozumienie, mimo że pan Dziadzio przedstawił bilans, można powiedzieć, wody i z tego wynikało, że Czesi sobie wykopali żwirownię, do której płynie woda i na dobrą sprawę to nie jest wina Turowa. Czas się kończy, więc mogę tylko powiedzieć, że chciałbym, żeby w Polsce była opozycja, która będzie stawać po stronie polskich interesów (Dzwonek), a nie po stronie interesów. Polskich interesów, nie rządu. A wy stajecie po stronie interesów każdego, kto na Polskę chce napaść i zrobić interes. Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Tomasz Piotr Nowak, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! To, co przed chwilą zaprezentował poseł Suski, to są po prostu pomówienia.

My jesteśmy polskimi patriotami i rozumiemy również interes energetyczny Polski. Dla nas kopalnia Turów jest czymś bardzo ważnym i powinna funkcjonować do końca lat 30., mówimy o tym w sposób zdecydowany. Propozycja stanowiska, którą zawarliśmy, właśnie tego dotyczyła - zobowiązania do skutecznych negocjacji przeprowadzonych przez premiera Morawieckiego z rządem czeskim w celu zabezpieczenia interesów i funkcjonowania kopalni Turów.

Nowelizacja ustawy o fotowoltaice będzie oparta jednak na funkcjonowaniu w obrocie handlowym, bo trzeba będzie sprzedać, prosument sprzeda energię po cenach hurtowych, a kupi ją po cenach detalicznych. W tym momencie dojdzie do obrotu handlowego, a projekty parasolowe, projekty z regionalnych programów operacyjnych, w które w tej chwili zaangażowanych jest dużo gmin i dużo mieszkańców tych gmin, mogą uzyskać dofinansowanie na poziomie 85%, wtedy kiedy nie ma handlowego aspektu.

Bardzo proszę, pan poseł Mieczysław Kasprzak, Koalicja Polska. Dziękuję bardzo. Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Po pierwsze, zablokowaliście wiatraki, a teraz mówicie, że będziecie budować na morzu dwa razy droższe. Blokowaliście fotowoltaikę na naszych dachach. W tej chwili jako wielki sukces ogłaszaliście przez kilka miesięcy to, co się stało. Polacy chcą inwestować w energię odnawialną, ale trzeba popatrzeć na to racjonalnie. Dzisiaj chcecie to wszystko zablokować, bo to, co pan opowiada, że się będzie rozwijać energia odnawialna prosumencka, jest nieprawdą.

Szkoda wam pieniędzy, żeby dać Polakom, żeby nawet mogli sobie zarobić, ale to jest racjonalne, bo pomagają państwu, inwestują własne środki finansowe. To, co chcecie w tej chwili zrobić, to będzie dramat. Po prostu chcecie zablokować rozwój energii odnawialnej. Rynek, ustawa mocowa - jest modyfikacja. To znaczy, że co? Że w dalszym ciągu wzrośnie obciążenie? Bo ja tak domniemywam i tak słyszałem. Prosiłbym bardzo o racjonalne podejście do tematu, bo rzeczywiście przez najbliższe lata całkowicie wyhamujecie zapał Polaków do tego, aby włączyć się w modernizację naszej energetyki. Uprzejmie dziękuję. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Bezpieczeństwo energetyczne Polski jest niewątpliwie związane z zieloną transformacją, z transformacją energetyczną. To jest droga, na którą powinniśmy wejść, i bardzo szybko nią podążać, ponieważ ona de facto oznacza suwerenność energetyczną, ona oznacza bezpieczeństwo energetyczne.

A kiedy słyszymy, że państwo zamierzają zmienić zasady rozliczeń energii, która jest pozyskana z fotowoltaiki, to tak, jakby do tego hamulca, który jest wciśnięty do podłogi, podnieść jeszcze ręczny do samego końca. Tak dzisiaj wygląda działanie rządu, jeżeli chodzi o transformację energetyczną, o wspieranie prosumentów, o wspieranie tej zielonej energii pozyskanej z natury. Pytanie do rządu. Czy rzeczywiście jest tak, że postanowiliście zahamować tę transformację energetyczną, zahamować wejście na drogę zielonej energii i po prostu nadal truć społeczeństwo paliwami kopalnymi? A społeczeństwo dzisiaj oczekuje zmiany. Społeczeństwo dzisiaj oczekuje, że będzie oddychało czystym powietrzem, że dzieci będą zdrowe, że nie będzie chorób, nie będzie umierało 50 tys. osób rocznie tylko dlatego, że mamy złe powietrze. Spali w kopalni. Chodzi o środowisko, chodzi o ludzi, którzy tam pracują, o twarz na arenie międzynarodowej i właśnie o przyszłość. Panie Ministrze! Dlatego chcielibyśmy wiedzieć, jaka jest strategia negocjacyjna. W jaki sposób zamierzacie rozmawiać z naszymi partnerami, bo to, co się dzisiaj dzieje, to jest po prostu absolutnie nieudolna (Dzwonek) próba przykrycia tego prowadzonego w sposób nieudolny tematu. Bardzo proszę, pan poseł Janusz Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni Państwo! Solidarna Polska broni suwerenności energetycznej Polski i broni przede wszystkim polskiego węgla, bo bez polskiego węgla nie ma taniej energii i nie będzie taniego ciepła. Niezrozumienie opozycji, która atakuje rząd, polega na tym, że nie rozumie jednej podstawowej rzeczy: za cenę energii i cenę ciepła, za ich wzrost odpowiada Unia Europejska, a więc unijny system handlu emisjami.

To dzisiaj Unia Europejska, a nie polski rząd hamuje transformację energetyczną.

A te pieniądze mogły być przeznaczone na inwestycje w nowe źródła energii, w niskoemisyjne źródła energii. To Unia Europejska i ten spekulacyjny mechanizm polega na tym, że w ciągu 7 lat, jeżeli dostaniemy z budżetu Unii Europejskiej 500 mld zł, to ponad 110, 120 mld zł polskie firmy będą musiały oddać Unii Europejskiej, do tego całego systemu właśnie na zakup uprawnień. Jakoby deficyt w tym całym systemie. To pokazuje, że to Unia Europejska doprowadza do tego, że będziemy płacić coraz więcej za energię i ciepło. Niestety w ciągu najbliższych miesięcy Polaków czekają ogromne podwyżki cen ciepła i energii. który prowadzi (Dzwonek) do tego, że Polska gospodarka jest coraz mniej konkurencyjna. Bardzo proszę, pan poseł Krzysztof Gadowski, Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze! Do roboty. Negocjować z Unią Europejską, walczyć o środki finansowe na transformację energetyczną, na to, o czym przed chwilą słyszeliśmy. Panie Ministrze! Pan mówił o programie „Mój prąd” Proszę nam powiedzieć, jak wygląda dziś „Mój prąd” Ile środków już jest przeznaczonych, ile Polacy czekają na te środki finansowe? Wspomniał pan o nowej ustawie. Wszyscy Polacy wiedzą, że waszą siłą sprawczą nigdy nie było to, żeby dążyć do rozwoju energetyki odnawialnej, energetyki związanej z OZE, z energią czystą i tanią. To nie była wasza mocna strona. Mało tego, zablokowaliście budowę energetyki wiatrowej na lądzie, a dzisiaj słyszymy o projekcie, o którym pan wspomniał. Państwo proponujecie zahamowanie rozwoju rozproszonej wielkiej elektrowni na dachach domów Polaków. Chcecie to zahamować. Mówicie, że ten system, który do tej pory funkcjonował, a był oparty na tym, że prosumenci produkują energię, nadwyżkę oddają do sieci i mogą odebrać 80% czy 70% tej energii za darmo, jest zły. Nie. To wszystko, ten system upustów jest zmieniamy na co? Na zwykłą sprzedaż. I w tym też nie byłoby nic złego. Ale wy mówicie znowu tak: energia, którą prosument będzie musiał kupić, kiedy jego elektrownia nie pracuje, będzie kosztowała dwukrotnie więcej niż sprzedana przez niego nadwyżka. Polacy wam po prostu już nie wierzą. To jest ten system. To jak to ma funkcjonować? Przeraziliście się kreatywności Polaków.

A wy dzisiaj mówicie, że nie. Po co te zmiany?

Bardzo proszę o przestrzeganie limitu czasu. Bardzo proszę, pan poseł Andrzej Szlachta, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, a właściwie dziesięcioleci, polski bilans energetyczny opierał się na paliwach kopalnianych. Dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął modernizację mocy wytwórczych oraz dywersyfikację struktury wytwarzania energii. Ponieważ dotychczasowy bilans energetyczny opierał się na paliwach kopalnianych, transformacja gospodarki do modelu niskoemisyjnego będzie wymagała dużych wysiłków społecznych, sektorów gospodarki i regionów, których funkcjonowanie w dużym stopniu wiąże się z wykorzystaniem wysokoemisyjnych paliw. Polski rząd planuje przeprowadzenie transformacji energetycznej w sposób ewolucyjny.

Wielkim wyzwaniem będzie poprawa efektywności energetycznej gospodarki.

Zwracam się do pana ministra z pytaniem: Jaki procent środków z Krajowego Programu Odbudowy zostanie skierowany na działania związane ogólnie z klimatem? Bardzo proszę, pani poseł Urszula Zielińska, Koalicja Obywatelska.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W ciągu tylko ostatnich 6 miesięcy na adres mojego biura poselskiego Ministerstwo Klimatu i Środowiska przysłało trzy pakiety książek i publikacji, materiałów promocyjnych. Wszystkie bez wyjątku promują energetykę jądrową. Mnie jako posłankę partii Zieloni, członkinię komisji energii i klimatu bardzo interesują sprawy transformacji energetycznej, redukowania emisji, więc z ochotą zabrałam się do lektury. A tam, proszę państwa, takie kwiatki. W rozdziale 11 zatytułowanym „Bez węgla nie ma światła” czytamy: Za mało naszych elektrowni przestawia się na węgiel, czyli to źródło energii, którego mamy najwięcej - Jimmy Carter.

Jaki był koszt tych publikacji? Czy Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi tak aktywną promocję, aż prosi się, żeby powiedzieć: lobbing, tylko na rzecz branży jądrowej czy również innych branż energetycznych? I w końcu: Dlaczego ministerstwo klimatu tak aktywnie promuje to jedno źródło energii? I wreszcie, panie ministrze, tak jak stabilny miks energetyczny wymaga przynajmniej kilku zróżnicowanych źródeł energii, tak i dobra edukacja i wiedza [[Dzwonek]] wymagają kilku źródeł informacji, więc w tym duchu pozwolę sobie przekazać bardzo dobrą publikację na ręce pana ministra. To jest książka autorstwa fizyka jądrowego Marcina Popkiewicza „Rewolucja energetyczna” Ona na s. 375 przedstawia, jak może wyglądać niskoemisyjny miks energetyczny, bezpieczny, stabilny dla Polski, bez węgla czy energii jądrowej w podstawie.

Bardzo proszę, pan poseł Jan Warzecha, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Czy w związku z transformacją energetyczną, z koniecznością osiągnięcia Europejskiego Zielonego Ładu, neutralności klimatycznej, z odejściem od węgla, dekarbonizacją zauważył pan minister zaangażowanie byłego przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, a obecnie przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej, w to, aby Polska nie poniosła ogromnych kosztów związanych z transformacją, czyli żeby cena energii nie wzrosła dla odbiorców indywidualnych i dla odbiorców przemysłowych? Drugie pytanie mam takie: Czy w związku ze wzrostem cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, a taki wzrost nastąpił w ciągu ostatniego roku z 25 euro do 50 euro. Jest dyrektywa, która wprawdzie w jakiś sposób redukuje ten wzrost, jednak ona okazuje się nieskuteczne, gdyż może być wdrożona wtedy, kiedy przez pół roku utrzymują się ceny trzykrotnie wyższe niż średnia cena uprawnień w ostatnich 2 latach.

Tu chciałem zapytać, czy rząd. Wiem, że rząd już podjął działania w tej mierze, żeby ten stan rzeczy zmienić, żeby ten mechanizm, który został wdrożony, zmienić na tyle, żeby zadziałał i żeby można było ograniczyć te wzrosty cen emisji do takich rozmiarów, jakie są w tej chwili. Bardzo proszę, pani poseł Małgorzata Chmiel, Koalicja Obywatelska. Dziękuję. Słuchając pana ministra, nie mogę się nadziwić, jak ten rząd dba o energię odnawialną, czyli nasze zdrowie.

W praktyce to ok. 2 km. Zasada działa również w drugą stronę, bo na terenie wokół tych elektrowni wiatrowych nie można budować. Wykluczone są więc duże połacie naszego terenu.

Obecnie 2% terytorium jest wyłączone z zabudowy mieszkaniowej w związku z tą ustawą, czyli to jest mniej więcej powierzchnia (Dzwonek) całego województwa opolskiego. Wójtowie, burmistrzowie zwracają się.

Bardzo proszę, pan poseł Grzegorz Lorek, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wracając jeszcze do Turowa, chciałem przypomnieć, że we wrześniu tego roku będzie zakończona budowa prewencyjnego ekranu chroniącego wody gruntowe na granicy kopalni. Dodatkowo zgodnie z trwającymi rozmowami planowana jest budowa wału ziemnego, który będzie zabezpieczał czeską stronę przed pyłami kopalnianymi.

Do tej pory zrealizowanych jest wiele inwestycji z myślą o mieszkańcach regionu, np. budowa ekranów akustycznych oraz instancji do zraszania ciągów węglowych czy też wymiana krążników w taśmociągach na cichobieżne, co sprawia, że kopalnia nie emituje tyle hałasu, ile było dotychczas.

Dziękuję. Bardzo proszę, pani poseł Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Mam wrażenie, że to, co wy nazywacie polityką energetyczną, to jest jakiś pomysł na sabotaż energetyczny. Przypomnę, że jak tylko doszliście do władzy, to pierwsza decyzja, którą podjęliście, dotyczyła kwestii związanej z elektrowniami wiatrowymi, czyli ograniczeniem energetyki wiatrowej w Polsce. I przypomnę, ponieważ ostatnio spotkał mnie jeden z parlamentarzystów, który powiedział coś takiego: zadałem pytanie o analizy związane z energetyką wiatrową, dlaczego zmieniono przepisy. Czyli nie wynikała ona z jakichś analiz, tylko wynikała po prostu z woli politycznej. W ten sposób oczywiście nie osiągnęliśmy celów, które były związane z energetyką, z OZE. Powiem więcej, jeżeli tu mówimy o płaceniu za emisję

Kolejna kwestia: Turów. Nieumiejętność rozmowy z Czechami. Doprowadziliście do sytuacji, w której zaraz możemy płacić kary w wysokości 5 mln euro dziennie. Awarie w Bełchatowie, nieumiejętności, zmiany kadrowe - efekt jaki mamy, taki mamy. Kwestia fotowoltaiki. Jak ludzie wreszcie wzięli sprawy w swoje ręce i postanowili zadbać o przyszłość swoich dzieci, o swoją kieszeń, ponieważ prąd jest drogi, to wy chcecie zrobić wszystko, żeby to też zabić. Zabiliście energetykę wiatrową (Dzwonek), chcecie zabić jeszcze fotowoltaikę. Dziękuję bardzo. Pani poseł Anna Ewa Cicholska, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę, pan poseł Piotr Borys, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek!

Otóż to, co wydarzyło się w ostatnim czasie, nie sprawia wrażenia, że państwo nad czymkolwiek panujecie.

Ale przede wszystkim Turów. Turów, w którym pracownicy elektrowni kopalni czekają na szybkie rozwiązanie sprawy. Turów, worek turoszowski, powiat zgorzelecki są podwójnie karane, po pierwsze, ogromnym zagrożeniem wynikającym z wyroku TSUE, groźbą codziennych kar, po drugie, brakiem szansy na sprawiedliwą transformację.

Państwo nie chcecie realizować tego projektu. Ten 1 mld zł przeznaczony na sprawiedliwą transformację - jego po prostu nie będzie, państwo z niego zrezygnowaliście w tym czasie. Nie mogę zgodzić się z tym, co wydarzyło się w Turowie. To jest ogromny zawód polskiej dyplomacji w tych wielomiesięcznych negocjacjach z Czechami. Już pomijam kwestię braku ambasadora. Po drugie, państwo nie potrafiliście, co wykazał także TSUE w swoim uzasadnieniu, przedstawić argumentów, w jaki sposób środek zapobiegawczy może zagrozić w kwestii funkcjonowania elektrowni i kopalni. Wprost wskazał to TSUE w swoim komunikacie. Muszę to przeczytać i proszę pana ministra o wycofanie tych skandalicznych słów, bo one nie wpływają korzystnie na możliwość negocjacji z Czechami. Przeczytam.

To piszą związkowcy. Apeluję, żeby to wycofali, i mówię to także do polskiego rządu i do pana ministra Sasina. Dziękuję bardzo. I bardzo proszę, pan poseł Marek Polak, Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma pana posła. Pan poseł Cezary Grabarczyk, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Pamięta pan, gdy ostatni raz był pan w Sejmie, rozmawialiśmy o awarii, która wyłączyła 10 bloków energetycznych w Bełchatowie. Tylko skończyliśmy, rozjechaliśmy się do domów i mieliśmy kolejną awarię związaną z pożarem. Pan kwestionował tezę, którą stawiałem wówczas, że w kopalni źle się dzieje, że nie ma właściwego nadzoru. Ten kolejny fakt potwierdził, że to ja miałem rację. Dziś mówimy o energetyce, o bezpieczeństwie energetycznym Polski w kontekście kłopotów w Turowie.

To pokazuje, że rząd kręci, że rząd oszukuje Polaków. Plan sprawiedliwej transformacji województwa łódzkiego nie ma żadnego umocowania w rozporządzeniu europejskim, ponieważ Bełchatów w tym rozporządzeniu nie jest ujęty.

Żadna z inwestycji realizowanych przez rząd PiS nie jest realizowana terminowo. Co będzie, gdy wyłączymy Bełchatów, a nie będzie jeszcze źródeł zastępczych?

Pani poseł Barbara Bartuś, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Debata, która odbywa się teraz w Sejmie, jest bardzo ważna, bo mówimy dzisiaj o bezpieczeństwie - o bezpieczeństwie energetycznym.

Proszę? Chcę powiedzieć, że w kontekście bezpieczeństwa energetycznego to, co państwo zrobiliście na moim terenie, ziemi gorlickiej, która była kolebką wydobycia ropy naftowej. Dzisiaj cieszymy się, że poparliście uchwałę o tym, że Nord Stream to jest coś złego, bo całe lata waszego funkcjonowania nie wskazywały na to, że działacie w interesie Polski. w Parlamencie Europejskim donosi na Polskę, chce, żeby Polsce zabrać pieniądze. jak opozycja walczy o to, żeby przedstawić Polskę w jak najgorszym świetle w TSUE. Padły tutaj słowa, które uważaliście za obraźliwe, słowa mojego kolegi, że tak się zachowują zdrajcy. Szanowni państwo, nie mówię tego, żeby atakować, ale zastanówmy się, w którym kierunku idziecie. Dużo złego stało się przez te 8 lat rządów, które mieliście. Dużo zostało w Polsce zniszczone, wyprzedane, zlikwidowane.

Dlatego apeluję o opamiętanie. Dziękuję, pani poseł. Ale ciągłe mówienie o opozycji, że nie są patriotami, i sugerowanie, że są zdrajcami, naprawdę nie jest na miejscu. Naprawdę uważam, że to lekka przesada, ponieważ jesteśmy wybrani przez Polaków, jesteśmy patriotami i mamy prawo i obowiązek być tutaj i mówić to, co uważamy za słuszne. Bardzo proszę, pan poseł Paweł Poncyljusz. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Ja to się dziwię, że pan jeszcze pracuje w tym ministerstwie, bo wszystkie kłopoty związane z Turowem to pana zasługa. Pan ignorował Czechów od kilku lat.

Ano to, że w pana ministerstwie zmieniono prawo odnośnie do oceny oddziaływania na środowisko.

Dlaczego pan tego nie napisał?

Pan jest za to osobiście odpowiedzialny.

Pan się po prostu do tego nie nadaje.

Dziękuję bardzo.

Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Padło tu już wiele różnych słów.

Też jestem za tym, żeby kopalnia Turów mogła funkcjonować. Ale tu niektórzy zapomnieli, że tuż po decyzji TSUE wielu przedstawicieli Platformy Obywatelskiej mówiło: tak, wyrok trzeba natychmiast wykonać.

No tak, oczywiście.

Program „Mój prąd” cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Jestem też oczywiście za odnawialnymi źródłami energii. Jednocześnie mam pytanie dotyczące ostatniej zimy. Mam pytanie związane z zakupem energii przez Szwecję. W związku z tym, że odnawialne źródła energii w czasie zimy nie wyprodukowały tyle prądu, ile powinny, nasz brudny prąd cieszył się dużym powodzeniem.

To wąskie gardło powoduje, że w tej chwili państwo tak naprawdę zmieniacie tę ustawę związaną z fotowoltaiką. Chcecie doprowadzić do tego, żeby ta fotowoltaika została ograniczona. Prawda jest taka, że mamy kłopoty.

Druga sprawa to Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Jak wiemy, on jest i będzie funkcjonował w najbliższych latach.

Słyszymy o Mysłowicach. Co w tym momencie? Czy może będzie tak, że nie sięgną po te pieniądze, w ogóle Śląsk nie sięgnie? To jest bardzo istotna sprawa.

Wydaje się, że oprócz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, pieniędzy z funduszy modernizacyjnych itd., powinno być takie działanie rządu, które będzie przyciągało w te rejony nowe inwestycje, np. dzięki specjalnym strefom ekonomicznym, które powinny działać na równych prawach na terenie całego kraju, a docierają głosy, że są równe i równiejsze.

Doliny wodorowe. Czy te doliny wodorowe będą związane z miejscem produkcji tego wodoru?

Elektrownia jądrowa.

A my do tej pory tak naprawdę nie mamy tych lokalizacji. Chciałbym w związku z tym zapytać: Kiedy ostatecznie rząd powie, że lokalizujemy pierwszą elektrownię na Pomorzu, drugą np. w Bełchatowie, a trzecią np. w Pątnowie? Czy taka kolejność jest i czy państwo już zdecydowaliście?

Sprawa ciepła - to jest fundamentalna sprawa - i modernizacji tych elektrociepłowni, które są elektrociepłowniami węglowymi.

W trybie sprostowania pan poseł Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość. To pan nie ma wiedzy. Odsyłam do mojego Facebooka, gdzie pokazałem, na czym polega luka unijnego systemu handlu emisjami. Bardzo krótko: 170 mln t uprawnień potrzebuje polska gospodarka, 105 mln t uprawnień mamy za darmo: 40 mln t uprawnień - instalacje, 65 mln - dla polskiego państwa na aukcje. 170 mln odjąć 105 mln to jest 65 mln - deficyt. Po prostu pan nie rozumie tego systemu. To oznacza, że te 65 mln t muszą polskie firmy kupić, płacą za to po 55 euro, i te pieniądze idą na giełdę w Lipsku, do Londynu, wypływają z Polski. nie ma problemu. To nie jest kwestia polityczna. Porozmawiajmy o tym. przede wszystkim ten system hamuje transformację energetyczną. Siądźmy, porozmawiajmy, wytłumaczę panu. Bardzo proszę o zabranie głosu podsekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska pana Piotra Dziadzię. Bardzo proszę, panie ministrze.

Szanowni Państwo!

Te projekty parasolowe będą elementami konsultacji publicznych i czekamy właśnie na tego typu uwagi od państwa i od prosumentów, od konsumentów.

Pytanie pana posła Kasprzaka.

Fotowoltaika nadal będzie systematycznie rozwijana. Nowe rozwiązania powodują to, że uzyskujemy na tych rachunkach nawet do 50% oszczędności.

Jeśli chodzi o ustawę mocową, to tutaj redukujemy obciążenia dla odbiorców o płaskim profilu zużycia i będziemy premiować tych, którzy nie powodują problemów w systemie. Taki jest cel też rynku mocy.

Jeśli chodzi o aukcje dla OZE, to w Sejmie jest projekt przedłużający te aukcje do 2027 r. Jeśli chodzi o pana posła Kowalskiego, to on już odpowiedział, wyjaśnił bardzo czytelnie sytuację związaną z ETS-ami - to jest prawda.

Dobrze, pan poseł Gadowski. Niedługo rozpocznie się trzecia edycja tego programu. To jest kolejne wsparcie dla prosumentów, to jest kolejne wsparcie dla rozwoju energetyki prosumenckiej. Jeśli ona nie będzie budowana w sposób odpowiedzialny, to w pewnym momencie nikt z tego nie będzie miał korzyści. Uważamy, że prosument będzie mógł również sprzedawać drożej wyprodukowaną energię elektryczną.

To prosument będzie decydował tak naprawdę o tym, jaka będzie cena.

Ten system, który w tej chwili jest budowany - prosumencki system - ma wykorzystać kreatywność Polaków, i wykorzystuje. W tym celu są te zmiany projektowane. Planujemy też w tym projekcie wspierać magazyny. Szanowni Państwo! Było powiedziane, że odbieramy prosumentom to, co daliśmy.

Jeśli chodzi o pytania pana posła Szlachty, jakie będziemy przygotowywać kluczowe projekty, które będą dotyczyły tak naprawdę efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Będziemy wykorzystywać zrównoważone i neutralne technologicznie odnawialne źródła energii. Będziemy rozwijać inteligentne systemy i sieci energetyczne oraz systemy magazynowania energii, w tym również magazynowania energii cieplnej. Będą inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie wodoru, magazynowanie, transport wodoru - to, o czym tak bardzo szeroko mówimy.

To jest dla nas zrozumiałe.

Jest gaz ziemny - też można go wykorzystywać w sposób ekologiczny poprzez systemy pozwalające na wyłapywanie dwutlenku węgla. Już są przygotowywane, mówiąc otwarcie. Jeśli chodzi o pana Jana Warzechę, jeśli chodzi o ETS, to oczywiście będziemy negocjować warunki w zakresie ETS-u, żeby te mechanizmy były bardziej sprawiedliwe. Kolejny element i kolejne pytanie to pytanie pana posła Chmiela. Były zarzuty, że likwidujemy zasadę 10H, ale niezależnie od tego, że ta zasada w jakikolwiek sposób ugrzęzła, wynikała ona tak naprawdę z dużych protestów w zakresie budowy energetyki wiatrowej.

Jeślibyśmy mieli informacje z czeskiej strony, moglibyśmy je realnie przeanalizować i realnie moglibyśmy zacząć rozmawiać. Więc, szanowni państwo, musi być równowaga, żebyśmy takimi danymi dysponowali i mówili. Warto go dokładnie przeanalizować, żeby zrozumieć, jak ten system pracuje.

Dobrze. Jeśli chodzi o sieci. Sieci oczywiście historycznie nie były zaprojektowane do takiej ilości odbioru i pan poseł doskonale z tego sobie zdaje sprawę.

To jest przewidziane i to się musi zrealizować. To tak szybko. W zasadzie to są chyba najważniejsze kwestie, które powinny zostać wspomniane.

Rynek mocy nie może finansować węgla. Będzie on w nowych aukcjach wspierał tylko źródła niskoemisyjne. I to w zasadzie chyba są te najważniejsze kwestie, które. Tak. Niskoemisyjne, przepraszam, niskoemisyjne, niegazowe.

Dziękuję bardzo, panie ministrze. Bardzo dziękuję. Wypowiedź ta kończy rozpatrywanie tego punktu porządku dziennego. Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich. Czy jeszcze ktoś z pań i panów posłów chce zgłosić się do wygłoszenia oświadczenia? Jeżeli nie, to zamykam listę. Bardzo proszę.

Wysoka Izbo! W moim wystąpieniu chciałbym poruszyć bardzo ważną kwestię ostatnich tygodni. Powiat, który bezpośrednio został dotknięty gradobiciem, powiat mi bardzo bliski, to powiat proszowicki, natomiast powiat sąsiadujący, czyli powiat krakowski również bardzo ucierpiał. Wiele gospodarstw potraciło swoje dochody, potraciło możliwości zarobkowania w tym roku. Problem jest poważny. Problem dotyczy ubezpieczeń. Problem poruszany już kilkanaście tygodni temu. Opozycja przyjechała na miejsce zdarzenia, również parlamentarzyści, których poprzednicy w 1992 r. mówili o tym, że ubezpieczenia w rolnictwie nie powinny być powszechne, powinny być dobrowolne; nie powinno być wspólnych ubezpieczeń, nie powinno być sytuacji, w której rolnicy w jakiś sposób mieliby się konsolidować, jeżeli chodzi o te ubezpieczenia.

Tak naprawdę od wszystkiego. Różnica polega na tym, że do końca nie wiemy, czy naszą uprawę zniszczy susza, grad czy deszcz nawalny. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć.

I dlatego 20 kwietnia tego roku złożyłem interpelację do ministra rolnictwa pana Grzegorza Pudy. Ta interpelacja spotkała się z pozytywnym odzewem, dlatego że pan minister obiecał w odpowiedzi poprzez swojego sekretarza stanu Ryszarda Bartosika, że w następnym roku dotowane ubezpieczenia dla rolnictwa będą priorytetem i kwoty zostaną podniesione. Natomiast jeżeli wystarczy pieniędzy z rezerwy budżetowej, na pewno rolnicy dostaną dodatkowe pieniądze. Chciałbym również podkreślić, że opozycja kłamała, że nie było reakcji Zjednoczonej Prawicy. Później w sytuacji, w której pan premier odwiedził Kraków razem z panem ministrem rolnictwa, udałem się na spotkanie z panem premierem i panem ministrem rolnictwa. Ta sytuacja dotyczyła prezentacji Nowego Ładu dla rolnictwa, Polskiego Ładu dla rolnictwa. Zasygnalizowałem właśnie o problemie w Małopolsce, jeżeli chodzi o ubezpieczenie, jeżeli chodzi o gradobicie. Wystosowałem interpelację do pana ministra rolnictwa, ponowną interpelację oraz do pana premiera Mateusza Morawieckiego w takiej kwestii, aby uruchomić tę rezerwę, aby pieniądze przekazać rolnikom, aby mogli skorzystać z tych pieniędzy dużo wcześniej, i aby zaplanować kolejny projekt, który by zapobiegał tego typu sytuacjom w przyszłości. Spotkałem się z pozytywnym odzewem. Pan premier obiecał, że prace na ten temat będą rozpoczęte, aby sytuacje związane z gradobiciem, ale nie tylko gradobiciem, ogólnie związane z trudnymi warunkami atmosferycznymi w rolnictwie, nie dotykały rolników w ten sposób, że rolnicy tracą dorobek życia poprzez to, że nie trafili z ubezpieczeniem od kataklizmu, że ubezpieczyli się od innych warunków atmosferycznych niż te, które akurat ich spotkały, od nieodpowiedniego kataklizmu. Bardzo serdecznie dziękuję za prace podjęte przez pana ministra Grzegorza Pudę oraz pana premiera Mateusza Morawieckiego. Cieszę się, że współpraca Zjednoczonej Prawicy w kontekście rolnictwa się układa. Są kolejne projekty wynikające z Polskiego Ładu, chociażby o podwykonawcach w rolnictwie, którzy nie płacą, załóżmy, pieniędzy rolnikom. Dziękuję ministrowi Zbigniewowi Ziobrze za reakcję w poprzedniej kadencji, kiedy odzyskaliśmy kilkanaście milionów dla rolników poszkodowanych przez firmy tytoniowe. Zjednoczona Prawica, droga opozycjo, dba o rolników. Bardzo proszę, pan poseł Mariusz Gosek, Prawo i Sprawiedliwość.

Wysoka Izbo! Chciałbym podziękować Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, na czele z panem ministrem Mariuszem Kamińskim, za stałe wsparcie jednostek ochotniczych straży pożarnych. Chciałbym także podziękować instytucjom rządowym, na czele z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, za to wsparcie. Jutro w regionie świętokrzyskim duże wydarzenie, mianowicie dojdzie do przekazania 30 wozów jednostkom ochotniczych straży pożarnych, pięć kolejnych wozów trafi do jednostek Państwowej Straży Pożarnej. 21 promes na kolejne dofinansowania trafi do 21 innych jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Często to strażacy - i to pokazują statystyki - są pierwsi na miejscu zdarzeń, wypadków drogowych, zdarzeń losowych. Była chęć, wola niesienia pomocy, ale brakowało profesjonalnego sprzętu. Tutaj z inicjatywą wyszły Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Fundusz Sprawiedliwości. Z tego miejsca chciałbym podziękować ministrowi sprawiedliwości, prokuratorowi generalnemu Zbigniewowi Ziobrze. Głęboko ufam, że one będą kontynuowane, bowiem wszyscy parlamentarzyści zapewne stoją na stanowisku, że wspieranie ochotników to też podnoszenie poziomu bezpieczeństwa Polaków, bezpieczeństwa podczas wszelkich akcji, w których druhowie ochotnicy uczestniczą. Raz jeszcze serdeczne podziękowania dla pana ministra Mariusza Kamińskiego i pana ministra Zbigniewa Ziobry za stałe wspieranie jednostek ochotniczych straży pożarnych. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Waldemar Andzel, Prawo i Sprawiedliwość.

Podczas II wojny światowej został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec, skąd uciekł, aby ponownie zaangażować się w działalność konspiracyjną.

Po ujawnieniu się był więziony 4 lata na zamku lubelskim za nieszczere ujawnienie się i ukrywanie czynów mjr. Dekutowskiego. Był szykanowany przez władze komunistyczne za przynależność do Armii Krajowej. Upamiętniał żołnierzy wyklętych, działał w Stowarzyszeniu Wolność i Niezawisłość oraz w stowarzyszeniu więźniów politycznych okresu komunistycznego. W 2020 r. Marian Pawełczak został awansowany na stopień pułkownika oraz odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Na tym zakończyliśmy oświadczenia poselskie. Informacja o wpływie interpelacji, zapytań oraz odpowiedzi na nie dostępna jest w Systemie Informacyjnym Sejmu. Protokół posiedzenia będzie wyłożony do przejrzenia w Sekretariacie Posiedzeń Sejmu.

Zamykam posiedzenie.